Otwieram posiedzenie.

Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Agatę Borowiec, Krzysztofa Truskolaskiego, Sylwestra Tułajewa i Monikę Wielichowską. W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Agata Borowiec i Sylwester Tułajew. Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Agata Borowiec i Monika Wielichowska. Protokół 59. posiedzenia Sejmu uważam za przyjęty wobec niewniesienia zastrzeżeń. Informuję, że na skutek wycofania przez wnioskodawców projektu uchwały w sprawie potępienia nazizmu, faszyzmu i komunizmu, zawartego w druku nr 2231, punkt porządku dziennego dotyczący tego projektu stał się bezprzedmiotowy. Na 59. posiedzeniu Sejm nie przeprowadził głosowań nad wnioskami o odrzucenie w pierwszych czytaniach poselskich projektów ustaw: - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, - o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Są to druki nr 2034, 2122 i 2182. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące te głosowania. Rada Ministrów przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Jest to druk nr 2334. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawiła opinię dotyczącą wniosku w sprawie wyboru uzupełniającego członka Trybunału Stanu, druk nr 2339. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tej sprawy. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, druk nr 2314. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o rządowych projektach ustaw: - o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym, - o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, - o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, - o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń. Są to druki nr 2278, 2308, 1928 i 2242. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę rozumiał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktu: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, druk nr 2291.

Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono wniosek o przeprowadzenie debaty nad sprawozdaniem komisji o uchwale Senatu w sprawie nowelizacji Prawa łowieckiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przeprowadzenie debaty nad sprawozdaniem o uchwale Senatu w sprawie Prawa łowieckiego, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm wniosek przyjął. Proponuję, aby Sejm wysłuchał w debacie. Proponuję, aby Sejm wysłuchał w debacie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Ktoś zgłasza sprzeciw, ale prosiłbym o to.

Został zgłoszony sprzeciw wobec 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

Kto z państwa posłów jest za przeprowadzeniem dyskusji oraz za wysłuchaniem 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Gdyby go nie przyjął, to wówczas mielibyśmy 5-minutowe.

Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm przeprowadził debatę średnią nad informacją ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 r. Prezydium Sejmu proponuje także, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusjach nad pozostałymi punktami porządku dziennego. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę rozumiał, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych przedłożyła sprawozdania: - w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz, zawarte w druku nr 2047, - w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika z dnia 12 września 2017 r. uzupełnionego w dniu 20 października 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru, zawarte w druku nr 2173, - w sprawie wniosku naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego, zawarte w druku nr 2306. Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec utrzymania w porządku dziennym tych sprawozdań. Są to, w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu, punkty sporne porządku dziennego. Propozycje utrzymania w porządku dziennym tych sprawozdań poddam kolejno pod głosowanie. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowania te nie są poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przystępujemy do głosowania nad sprawozdaniem komisji dotyczącym pani poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz. Kto z państwa posłów jest za utrzymaniem w porządku dziennym punktu: sprawozdanie komisji dotyczące immunitetu pani poseł, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad sprawozdaniem komisji dotyczącym posła Ryszarda Petru. Kto z państwa posłów jest za utrzymaniem w porządku dziennym punktu: sprawozdanie komisji regulaminowej dotyczące immunitetu pana posła Ryszarda Petru, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm propozycję przyjął. Przystępujemy do głosowania nad sprawozdaniem komisji dotyczącym posła Stanisława Gawłowskiego. Kto z państwa posłów jest za utrzymaniem w porządku dziennym punktu: sprawozdanie komisji regulaminowej dotyczące immunitetu, wyrażenia zgody przez Sejm na zatrzymanie posła Gawłowskiego, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm propozycję przyjął. Przypominam, że kluby złożyły wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o punkty: - Informacja prezesa Rady Ministrów na temat ustaleń poczynionych w trakcie analizy zapisów wideo i innych materiałów dokumentujących niezgodne z prawem zachowania uczestników i organizatorów Marszu Niepodległości, które polegały na propagowaniu faszyzmu, nawoływaniu do nienawiści na tle rasowym oraz publicznym znieważeniu grupy ludności ze względu na jej przynależność rasową - jest to wniosek zgłoszony przez Klub Poselski Nowoczesna, - Informacja prezesa Rady Ministrów na temat przyczyn porażki rządu Prawa i Sprawiedliwości w staraniach o przeniesienie siedzib Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) i Europejskiej Agencji Leków (EMA) z Londynu do Warszawy - zgłoszony przez Klub Poselski Nowoczesna, Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie godzących w wolność słowa oraz będących próbą zastraszenia działań policji oraz prokuratury wymierzonych przeciwko: - dziennikarzowi Wojciechowi Bojanowskiemu, który działając w interesie społecznym, obnażył patologię działania prokuratury oraz ujawnił rażące nadużycia policjantów na komisariacie Wrocław-Stare Miasto, którzy przekraczając swoje uprawnienia, mogli przyczynić się do śmierci Igora Stachowiaka, oraz: - dziennikarzowi Tomaszowi Piątkowi, autorowi książki „Macierewicz i jego tajemnice”, w której ujawnia powiązania obecnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza z byłymi agentami komunistycznej bezpieki oraz organizacjami mafijnymi wywodzącymi się ze służb specjalnych ZSRR - zgłoszony przez Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska. W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam kolejno pod głosowanie wnioski o uzupełnienie porządku dziennego.

Wysoka Izbo! Bardzo chętnie byśmy poparli ten wniosek, ale on musi być inaczej sformułowany.

Wtedy - chętnie - będziemy w stanie to poprzeć.

No nie jesteśmy w stanie zmienić tego wniosku. Proszę państwa, teraz możemy tylko to przegłosować. To jest wniosek klubu Nowoczesna. Klubu Nowoczesna nie widzę, nie słyszę. W związku z tym.

Kto z państwa posłów jest za ogłoszeniem przerwy, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek o przerwę odrzucił.

Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o ten punkt, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji w sprawie przeniesienia siedzib urzędów europejskich - wcześniej cytowałem, przedstawiałem cały tytuł wniosku. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o ten punkt, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji w sprawie działań policji oraz prokuratury dotyczących dziennikarzy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o ten punkt, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Informuję, że Konwent Seniorów jednomyślnie zaopiniował propozycję rozpatrzenia na bieżącym posiedzeniu informacji w sprawie osób odbywających kary pozbawienia wolności oraz wobec których zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze lub tymczasowe aresztowania, a które zostały uniewinnione w toku procesu lub w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji, a także w sprawie zadośćuczynień za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, o której przedstawienie wnosił Klub Poselski Kukiz’15. Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Informacja w tej sprawie, a także wykaz ustaw, które Senat przyjął bez poprawek, dostępne są w Systemie Informacyjnym Sejmu. Proszę pana posła sekretarza o odczytanie komunikatów. Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji: - do Spraw Petycji - godz. 10.15,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 Infrastruktury wspólnie z Komisją Finansów Publicznych - godz. 14.30, Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - godz. 15, - Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 15, - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 15, - Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 15, - Administracji i Spraw Wewnętrznych - godz. 16, - Obrony Narodowej - godz. 16, - Finansów Publicznych - godz. 17, - Infrastruktury - godz. 17, - Spraw Zagranicznych - godz. 18, - Obrony Narodowej - godz. 19. Dodatkowo informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych: - wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej i Parlamentarnego Zespołu ds. Energetycznego Pakietu Zimowego - godz. 14, - Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego - godz. 14, - Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju drobiarstwa jako strategicznej gałęzi polskiej gospodarki - godz. 16, - Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców „Polski powiatowo-gminnej” - godz. 16.30. Dodatkowo informuję, że duszpasterstwo parlamentarzystów serdecznie zaprasza panie i panów posłów na rekolekcje wielkopostne, które odbędą się w dniach od 21 do 23 marca br.

Rekolekcje poprowadzi ks. prof. Marek Kotyński z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Dziękuję. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (druki nr 2263 i 2278) Proszę panią poseł Alicję Kaczorowską o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić państwu sprawozdanie z pierwszego czytania, z rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie, rozpatrzyła ten projekt. W czasie procedowania przyjęto poprawki legislacyjne oraz doprecyzowujące i redakcyjne. Wszystkie one, w liczbie trzech, dotyczyły art. 2.

Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko co do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym z druków nr 2263 i 2278. Niniejszy projekt ma na celu usunięcie barier w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, w tym obejmujących budowę tuneli kolejowych, a także poprawę uregulowań dotyczących funkcjonowania kolei o charakterze historycznym i turystycznym. Wprowadzane zmiany są wynikiem postulatów podmiotów realizujących inwestycje na kolei, organizacji pozarządowych zrzeszających miłośników kolejnictwa. Organizacje pozarządowe od wielu lat postulowały wprowadzenie możliwości nieodpłatnego przekazywania mienia kolejowego. Projektowane rozwiązania będą stanowiły instrument wsparcia rozwoju i utrzymania historycznych i turystycznych linii kolejowych. Jednocześnie pozwolą one największym spółkom kolejowym na pozbycie się mienia, które jest zbędne do prowadzenia działalności, natomiast generuje tylko dodatkowe koszty. Zmiany w ustawie o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” obejmują m.in. wprowadzenie możliwości nieodpłatnego przekazania na rzecz organizacji pozarządowych mienia ruchomego PKP stanowiącego zabytki techniki kolejowej oraz materiałów odzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac remontowych lub modernizacyjnych. Zmiany ustawy o transporcie kolejowym przewidują nowe wyłączenie spod działania przepisów ustawy dla transportu kolejowego wykonywanego na liniach o szerokości toru poniżej 300 mm, co jasno ureguluje sytuację kolejek parkowych czy ogrodowych. Wprowadzone zmiany umożliwią zarządcom kolei wąskotorowych pozyskiwanie dofinansowania, w tym również ze strony zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. Obecna wersja przepisów wprowadza ułatwienia w eksploatacji czynnych pojazdów historycznych, którym nadano nową definicję. Odnośnie do inwestycji wymagających budowy tunelu w projekcie ustawy proponowane jest doprecyzowanie przepisów umożliwiających ograniczenie korzystania z nieruchomości. Ograniczenie to wprowadzone będzie w drodze decyzji wojewody wraz z udzielonym zezwoleniem na budowę lub przebudowę tunelu z infrastrukturą towarzyszącą. Zmiana ta pozwoli na prowadzenie działań inwestycyjnych oraz utrzymaniowych bez konieczności wykupu gruntów, pod którymi przebiega budowana infrastruktura. Prawa właścicieli, użytkowników lub posiadaczy gruntów zostaną zabezpieczone poprzez ustalenie prawa do odszkodowania z tytułu ustalonego ograniczenia własności. Rozwiązanie to ułatwi realizację inwestycji związanych z budową i modernizacją tuneli kolejowych, a także ich użytkowanie, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, gdzie w ramach realizacji ww. inwestycji można znacznie ograniczyć koszty związane z wykupem gruntów, problemy z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego, problemy z negatywnym oddziaływaniem na środowisko i bezpieczeństwo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ze względu na liczne pozytywne aspekty przedstawionych zmian Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie popierał rządowy projekt ustawy. Teraz głos zabierze pan poseł Cezary Grabarczyk w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym, druk nr 2263, zawiera szereg ciekawych rozwiązań. Pierwsza grupa przepisów dotyczy możliwości przekazywania linii kolejowych na rzecz samorządów. Dotyczy to całych linii, ale także odcinków linii kolejowych. Pod jednym wszakże warunkiem: w celu dalszej eksploatacji tych linii na czas nie dłuższy niż 3 lata. Zarządca tych linii będzie mógł przekazywać linie do dalszej eksploatacji bez zgody ministra infrastruktury. To ułatwi podejmowanie decyzji. Druga grupa przepisów dotyczy możliwości przekazania majątku spółki PKP lub innych spółek kolejowych na rzecz organizacji pozarządowych. Dotyczy to zarówno pojazdów o znaczeniu historycznym, jak i części linii kolejowych, urządzeń, które są efektem odzyskanym przy remontach, modernizacji linii kolejowych. Beneficjentem mogą być nie tylko organizacje pozarządowe, ale także samorząd - choćby ten samorząd, który przejął do dalszej eksploatacji część linii kolejowych bądź też całą linię kolejową. Na podkreślenie zasługuje sprecyzowanie katalogu warunków, które muszą spełnić beneficjenci. Te rozwiązania mogą pozwolić nie tylko na zmniejszenie kosztów spółek kolejowych, ale także na zwiększenie atrakcyjności turystycznej małych ojczyzn. To jest dobre rozwiązanie, zasługuje na poparcie. Ale fundamentalna zmiana dotyczy możliwości ograniczenia własności w związku z planowanymi inwestycjami, które wymagają drążenia tunelu. I na te rozwiązania tak naprawdę czekają wykonawcy, którzy już podpisali umowę na budowę tunelu kolejowego w Łodzi między dworcem Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska. Oni tak naprawdę nie mają dzisiaj możliwości rozpoczęcia realizacji tej inwestycji, bo nad tymi przepisami dopiero w tej chwili procedujemy. Te przepisy zasługują na poparcie. Dlatego klub Platformy Obywatelskiej poprze te rozwiązania. Warto przy tej okazji zapytać, czy nie należałoby pójść jeszcze dalej, bo w Ministerstwie Infrastruktury trwały już prace nad rozwiązaniami, które dotyczyłyby prawa zabudowy - podobne prace trwały w Ministerstwie Sprawiedliwości - bądź też tzw. własności warstwowej, inaczej też określanej jako własność 3D. Dlaczego? Dlatego że proponowane rozwiązania, które powodują ograniczenie prawa własności na potrzeby realizacji inwestycji tunelowych, rozwiązują tylko część problemów, ale przede wszystkim nie uwalniają gigantycznego potencjału, który drzemie w nieruchomościach zajętych przez linie kolejowe przebiegające w obrębie wielkich miast, w obrębie [[Dzwonek]] aglomeracji. które dotyczą własności warstwowej, pomogłyby uruchomić ten potencjał. Jest pan poseł?

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Europejskich Demokratów pragnę przedstawić stanowisko, uwagi co do sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, zawartych w drukach nr 2263 i 2278. Jak możemy wywnioskować i jak czytamy w projekcie rządowym, jak i według tego, o czym mówiliśmy na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, projekt dotyczy, można powiedzieć, ułatwienia funkcjonowania kolei i usunięcia barier przez uzupełnienie i doprecyzowanie obecnych uregulowań w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, w tym obejmujących m.in. budowę tuneli kolejowych, a także uregulowań dotyczących funkcjonowania kolei o charakterze historycznym i turystycznym.

W części pierwszej mówimy o inwestycjach, o zmianie formuły realizacji inwestycji. Wymaga to działań związanych z szeroko rozumianymi regulacjami stanów prawnych, ale w założeniu, taki jest cel, ma to doprowadzić do ułatwienia przygotowania, spełnienia wymogów, które poprzedzają sam moment rozpoczęcia inwestycji, a dalej - również eksploatacji i utrzymania całości infrastruktury kolejowej w kolejnych latach.

Najczęściej mamy tu na uwadze środki pochodzące z programów w obecnym okresie realizacji, jak również z programów zarządzanych na szczeblu krajowym, a niejednokrotnie dotyczy to również programów wdrażanych na poziomie regionów. W drugiej części mówimy o uproszczeniach, które mają dotyczyć tzw. pojazdów historycznych i infrastruktury, która służyła nam w minionym czasie.

Tak że klub będzie za kontynuowaniem tych prac i w nieodległym, stosownym czasie, po przygotowaniu, sfinalizowaniem i przyjęciem ustawy. Teraz pan poseł Mirosław Suchoń, klub Nowoczesna. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Szanowni Państwo! Projekt ustawy będący przedmiotem dzisiejszych obrad ma na celu wprowadzenie ułatwień w funkcjonowaniu kolei oraz usunięcie pewnych barier w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, w tym dotyczących budowy tuneli kolejowych. Projekt zawiera również propozycję nowych uregulowań dotyczących funkcjonowania kolei o charakterze historycznym i turystycznym. Z przedstawionego przez rząd uzasadnienia wynika, iż proponowane zmiany są wynikiem postulatów podmiotów realizujących inwestycje na liniach kolejowych, organizacji pozarządowych zrzeszających miłośników kolejnictwa, w szczególności formułowanych w trakcie prac zespołu do spraw ochrony zabytków kolejnictwa działającego przy senackiej Komisji Infrastruktury w okresie od lutego do sierpnia 2016 r. W odniesieniu do ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych, które już od wielu lat postulowały wprowadzenie możliwości nieodpłatnego pozyskiwania mienia kolejowego. Rozwiązania zawarte w projekcie mogą ułatwić prowadzenie działalności statutowych i o charakterze historycznym, w tym pozyskiwanie zabytków kolejnictwa i sprawowanie nad nimi opieki. Rozwiązania te mogą również stanowić instrument wsparcia rozwoju i utrzymywania historycznych i turystycznych linii kolejowych. Ponadto spółki kolejowe na podstawie projektowanych przepisów będą mogły przekazywać nieużytkowane mienie. To pewnego rodzaju ułatwienie, które pozwoli spółkom kolejowym na redukcję kosztów. Otwarte pozostaje pytanie, dlaczego z grona uprawnionych do nieodpłatnego przeniesienia linii kolejowej lub odcinka takiej linii w zarządzanie rząd wykreślił wskazanego wprost przedsiębiorcę, który musiał być wskazany przez jednostkę samorządu terytorialnego. Pomimo argumentów przedstawianych przez przedstawiciela rządu aktualne pozostaje pytanie, czy zmiany nie powinny iść jednak w kierunku poszerzenia uprawnień takich przedsiębiorców. Projekt wprowadza również szereg zmian w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Na uwagę zasługują m.in. przepisy dotyczące wprowadzenia wyłączeń w obowiązujących przepisach dla transportu kolejowego wykonywanego na liniach o szerokości toru poniżej 300 mm, co spowoduje lepsze uregulowanie sytuacji kolejek parkowych czy ogrodowych. Projekt wprowadza również nowe uregulowania, które umożliwią zarządcom kolei wąskotorowych pozyskiwanie dofinansowania z nowych źródeł, w tym również ze strony zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu kolejki będące często lokalnymi atrakcjami będą mogły lepiej wykorzystywać swój potencjał. W przedłożeniu przewidziano także rezygnację z dotychczasowego wyłączenia przepisów ustawy do pojazdów historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej. Oznacza to, iż wyłączenia te będą stosowane również do pojazdów poruszających się po sieci kolejowej. To rodzi pytania o kwestie bezpieczeństwa, ale mamy nadzieję, że rząd na to zadowalająco odpowie. Zmiany proponowane w przedłożeniu dotyczą również procesów inwestycyjnych na liniach kolejowych, może nawet przede wszystkim. W uzasadnieniu tych zmian rząd wskazuje, iż po ich wprowadzeniu znikną pewne bariery w prowadzeniu inwestycji kolejowych obejmujących budowę lub przebudowę tunelu oraz że zagwarantują one prawo do wejścia na teren nieruchomości, a także do dokonania prac związanych z konserwacją, utrzymaniem sieci lub usuwaniem awarii. Ponadto projekt zawiera rozwiązania dotyczące wywłaszczania i ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budownictwo kolejowe oraz zmiany dotyczące odstępstw od stosowania obowiązku technicznych specyfikacji interoperacyjności. Proponowane zmiany mogą spowodować, iż inwestycje kolejowe będą realizowane sprawniej i bardziej terminowo. To jest oczywiście odpowiedź na postulaty przedsiębiorców, którzy bardzo często mają problemy w tych obszarach. Należy jednak zauważyć, panie ministrze, że same przepisy nie wystarczą, trzeba profesjonalnego podejścia.

Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałbym przedstawić stanowisko Koła Poselskiego Wolni i Solidarni dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 8 września 2000 r. dotyczące przede wszystkim uregulowań w sprawie realizacji projektów inwestycyjnych i regulacji dotyczących funkcjonowania kolei o charakterze historycznym i turystycznym.

Te rozwiązania pozwolą na realizację projektu w zakresie modernizacji krajowej infrastruktury kolejowej, a tym samym na właściwe wykorzystanie środków finansowych funduszy Unii Europejskiej. Do tej pory mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której nie było możliwe nieodpłatne przejęcie linii kolejowej lub jej odcinka w zarządzanie przez przedsiębiorcę wskazanego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wprowadzone zmiany dopuszczą sytuację, w której jednostka samorządu terytorialnego może realizować funkcję zarządcy infrastruktury kolejowej, np. w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych. Proponowane zmiany będą korzystne także dla organizacji zajmujących się historią. Stowarzyszenia i fundacje będą mogły zostawać właścicielami zabytków kolejnictwa, będą mogły sprawować nad nimi opiekę, co również będzie stanowiło instrument wsparcia rozwoju i utrzymania historycznych i turystycznych linii kolejowych. Jednocześnie pozwoli PKP SA, PKP PLK SA na pozbycie się mienia, które nie jest obecnie wykorzystywane do prowadzenia ich bieżącej działalności. Przedmiotowa ustawa wprowadza pojęcie pojazdu historycznego i pojazdu turystycznego.

Dodanie w art. 4 w pkt 6i wyżej wspomnianej definicji ma na celu dookreślenie kategorii pojazdów użytkowych nie w celu zaspokojenia publicznych potrzeb transportowych, ale przede wszystkim zaspokajania potrzeb społecznych o charakterze np. emocjonalnym, związanych z pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego w danym regionie, edukacją techniczną, aktywnym spędzaniem czasu wolnego, turystyką infrastrukturalną, industrialną. Tak więc to jest charakter tego artykułu.

Zapisy te mają na celu uregulowanie kwestii związanych z budową tuneli w ramach inwestycji i projektów kolejowych. Doprecyzowano dotychczasowe normy, aby w sposób jednoznaczny i bezsporny wskazać na możliwość realizacji tych inwestycji. Uregulowanie kwestii związanych z realizacją projektów inwestycyjnych wymagających budowy tuneli jest szczególnie istotne w przypadku realizacji inwestycji liniowych prowadzonych w terenie zurbanizowanym, gdzie istnieją techniczne możliwości posadowienia inwestycji pod powierzchnią gruntu, bez konieczności dokonywania wywłaszczenia nieruchomości. W związku z pozytywnymi zmianami, jakie zaproponowano, Koło Poselskie Wolni i Solidarni poprze rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do pytań zapisało się sześcioro pań i panów posłów.

Jako pierwszy - pan poseł Zbigniew Gryglas, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Projektowana ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” to potrzebna i oczekiwana regulacja. Ułatwi ona restrukturyzację i właściwe wykorzystanie majątku kolejowego.

Bo to dopuszcza ustawa. I druga kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę - któryś z moich poprzedników już o tym mówił - to sprawa ustawy o własności warstwowej. To rzeczywiście bardzo potrzebna regulacja. Czy ministerstwo [[Dzwonek]] pracuje nad tą regulacją?

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pierwsze: Czy jesteście państwo przekonani, że te zapisy rzeczywiście spowodują pewne przyspieszenie, jeśli chodzi o realizację inwestycji na kolejach? Pytam, dlatego że wszyscy mamy świadomość, że te obsunięcia w realizacji projektów są bardzo duże.

I drugie pytanie: Czy zapisy dotyczące kolei wąskotorowych, tych historycznych czy tam parkowych, są wynikiem apeli i sugestii ze strony właśnie zarządców tych kolei, czy to państwo odgórnie uznaliście, że takie rozwiązania będą najbardziej korzystne? Pan poseł Cezary Grabarczyk, klub Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ustawa tunelowa rozwiąże ten jeden problem, jak drążyć tunele w warunkach wielkich aglomeracji, jak realizować linie kolejowe w tych tunelach, jak naprawiać, remontować je w przypadku uszkodzeń i awarii. Ale w wielkich miastach linie kolejowe przebiegają często przez sam środek, przez centra tych miast, często rozcinając miasta na części.

Bardzo proszę. Panie Ministrze!

A z drugiej strony czy wprowadzenie tej ustawy w jakikolwiek sposób może zaburzyć ten czas projektowania tuneli w Łodzi, czyli połączenie między Łodzią Kaliską a Łodzią Fabryczną? Pani poseł Zofia Czernow, klub Platforma Obywatelska. Panie Marszałku!

Ta bardzo piękna linia kolejowa, przebiegająca przez parki krajobrazowe, jest od 2 lat nieczynna. Mieszkańcy bardzo cierpią z tego powodu, można nawet mówić o wykluczeniu komunikacyjnym. Czy ta ustawa da szansę, aby szybciej przekazać tę linię do urzędu, do samorządu wojewódzkiego, który wyraża zgodę na jej przyjęcie i wyremontowanie? W odpowiedziach cały czas mnoży się bardzo wysokie koszty remontu, które chyba już wielokrotnie zostały na papierze zwiększone, a mieszkańcy cierpią. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, klub Nowoczesna. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jest wiele takich linii kolejowych, które wymagają remontów.

Panie Ministrze! Ja też poproszę o wyjaśnienia kwestii dotyczącej tego, kiedy, bo pan minister Grabarczyk słusznie tutaj pyta nie o to, czy ta ustawa dotycząca własności warstwowej pojawi się, ale kiedy ona się pojawi, bo rzeczywiście mogłoby to rozwiązać wiele problemów. Może warto podać przykłady linii turystycznych, historycznych, które na tych przepisach zyskają.

Zamykam listę posłów zapisanych do głosu. Teraz proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana Andrzeja Bittela. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W pierwszych słowach chciałem podziękować za tę dobrą ocenę przedłożenia rządowego, które dzisiaj mamy szansę omawiać. Postaram się w kilku słowach odnieść się do zadanych pytań i wątpliwości, które powstały na jego tle.

W związku z tym formuła pozostaje taka sama, a samorząd jest dla nas partnerem bardzo pewnym, tj. takim, na którym można polegać, który ma doskonale rozpoznane potrzeby społeczne - najlepiej. To chyba oczywiste na tej sali, że idea samorządności jest bardzo dobrym rozwiązaniem, i nie trzeba tego dłużej uzasadniać. Stąd też odwoływanie się do samorządu, a nie do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą - i bardzo dobrze, że taką prowadzą - ma inne cele. Samorząd ma na celu zaspokajanie potrzeb zbiorowych, a przedsiębiorcy mają na celu zarobkowanie i ta synergia spotka się dzięki tym przepisom. Pan poseł Meysztowicz zapytał, czy to rzeczywiście przyspieszy.

Pierwszy etap, czyli etap pozyskiwania nieruchomości i uzyskiwania tytułów prawnych w tym zakresie, jest zawsze skomplikowany, trudny, a odszkodowanie, słuszne odszkodowanie, które się należy właścicielowi, który albo ma ograniczone prawa, albo wręcz jest wyzuty z własności. Jest niezwykle ważne, żeby dla niego te przepisy były jasne, czytelne i na dodatek żeby procedury postępowały sprawnie.

Nie chciałbym wymieniać w tym miejscu i momencie linii kolejowych, które będą przyjmowane przez samorząd, które dzięki tej ustawie uzyskają wsparcie samorządu czy którym będzie łatwiej funkcjonować, bo takich przykładów jest naprawdę bardzo dużo.

To jest ogólny postulat - postulat, który się rodził, był powtarzany od lat. Wychodzimy naprzeciw potrzebom podmiotów, które prowadzą swoją stowarzyszeniową działalność w taki sposób, żeby pielęgnować tradycję kolejową, którą chcemy pielęgnować i która powinna być pielęgnowana tak, żeby udzielać wsparcia, tj. starać się mniej przeszkadzać, a więcej udzielać wsparcia.

Pan poseł Suchoń wspominał, że czas rozliczania już się podobno skończył.

Na poziomie Ministerstwa Infrastruktury rozważamy podjęcie takiej inicjatywy, bo mamy ogromne przeświadczenie o tym, że nawet z punktu widzenia ściśle sektorowego, kolejowego, takie rozwiązanie byłoby niezwykle pożyteczne z wielu różnych względów, również tych, które wymieniał pan poseł Grabarczyk.

Muszę to wyraźnie powiedzieć, żeby to wyraźnie wybrzmiało: sytuacja, w której znajdujemy się w ramach realizacji perspektywy bieżącej, europejskiej perspektywy bieżącej, w porównaniu do początku roku 2016 jest diametralnie inna.

Proszę mieć świadomość, że my w tej chwili, jak dobrze pójdzie, będziemy kończyli przetarg, który się toczy od połowy roku 2015, na GSM-R. A więc ten wysiłek, który został wykonany przez 2 lata przez beneficjenta, Polskie Linie Kolejowe, należy doceniać, należy go odbierać pozytywnie.

Tak więc chciałbym tu mocno powiedzieć, że postęp wykonany przez te ostatnie 2 lata jest ogromny. Dodatkowo dwa zdania.

być do niej znakomicie przygotowani. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2156 i 2308) Proszę pana posła Bogdana Rzońcę o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Ministrze!

Komisje: Finansów Publicznych i Infrastruktury przepracowały projekt artykuł po artykule.

Wpłyną one bezpośrednio na zmniejszenie obciążeń administracyjnych po stronie przedsiębiorców. Mając na uwadze różnice przy wykonywaniu przewozów drogowych i kolejowych, w projektowanej regulacji uwzględniono specyfikę przewozu koleją.

Proszę państwa, pomimo że zakazany jest wywóz za granicę leków zagrożonych brakiem dostępności w Polsce, problem nie został całkowicie rozwiązany i polskie apteki ciągle borykają się z problemem dostępu do innowacyjnych lub zaawansowanych leków. W związku z powyższym niezbędne jest objęcie systemem monitorowania przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych określonych właśnie w tej ustawie.

Na przykład w zmianie 3. był użyty termin „przemieszczenie”, natomiast po dyskusji zmieniono ten termin na „przemieszczanie” towarów.

A więc ten przepis zmienia tę sytuację.

Jest to konsekwencja wcześniejszych zmian.

Także w art. 16, proszę państwa, został zmieniony sens poprawki, który polega na tym, że w przypadku zajęcia przez inspekcję farmaceutyczną nielegalnie przewożonych leków będzie możliwe ponowne ich wprowadzenie do obrotu poprzez sprzedaż przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca przechowywania zatrzymanego towaru. Ma to służyć temu, aby deficytowe leki zagrożone wywozem nie czekały do końca postępowania - mogłyby się po prostu przeterminować - tylko od razu mogły zostać sprzedane i wprowadzone do obrotu. Celem takiego działania jest po prostu wzrost poziomu bezpieczeństwa lekowego państwa. Jeśli chodzi np. o poprawkę 5., która została zgłoszona, to ta poprawka wyłącza możliwość wstrzymania przez sąd administracyjny wykonania decyzji wydanej przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej w sytuacji, kiedy apteka lub hurtowania uczestniczyły w tzw. odwróconym łańcuchu dostaw i przyczyniły się do braku leczniczych produktów na polskim rynku. Obecnie każda decyzja organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jest wstrzymywana przez sąd administracyjny i nie podlega wykonaniu do czasu wydania prawomocnego wyroku sądu. Tymczasem właśnie taka sytuacja sprawia, że podmioty trudniące się nielegalnym wywozem leków z naszego kraju doskonale funkcjonują przez lata, bo sąd administracyjny po prostu wstrzymał decyzję Państwowego Inspektora Farmaceutycznego. A więc zmieniamy tę sytuację.

Tych zadań nie mogą wykonywać pracownicy korpusu służby cywilnej.

I ta poprawka wyraźnie mówi, precyzuje, że kontrola drogowa jest wyłącznie domeną funkcjonariuszy, a wszystkie pozostałe zadania związane z orzecznictwem mogą być wykonywane tylko przez cywilnych pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Ta poprawka jest kluczowa, ponieważ umożliwi ona współpracę Krajowej Administracji Skarbowej z ministrem zdrowia w zakresie skutecznej walki z nielegalnym wywozem leków w Polsce.

Proponuję Wysokiej Izbie jej przyjęcie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Pierwsza zabierze głos pani poseł Gabriela Masłowska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Chciałabym wobec tego zwrócić uwagę na kilka kwestii. Pragnę podkreślić, że nadrzędnym celem przedłożonego projektu ustawy jest walka z nadużyciami podatkowymi oraz przeciwdziałanie masowej sprzedaży produktów leczniczych przez hurtownie do zagranicznych kontrahentów kosztem polskiego rynku leków. Wprowadzenie w 2017 r. ustawy o monitorowaniu systemu drogowego przewozu towarów spowodowało, że przewóz towarów wrażliwych przeniósł się na środki transportu kolejowego, co potwierdza analiza Krajowej Administracji Skarbowej. Wymaga wobec tego objęcia nadzorem na wzór systemu drogowego uwzględniającym specyfikę kolei, także transportu kolejowego, co czynimy niniejszym projektem ustawy. Kwestia wywozu leków jest problematyczna, ponieważ powoduje brak leków w Polsce, zwłaszcza takich, które są istotne dla ratowania życia, nowoczesne, niezbędne. One są niedostępne dla polskich pacjentów. W związku z tym już od 2012 r. ten problem był monitorowany i zauważany, jednak cały czas jest nierozwiązany, narasta.

Część tych leków sprzedaje się na czarnym rynku bez opodatkowania VAT-em, CIT-em, PIT-em.

Chcemy z tym procederem podjąć walkę.

Dostosowanie systemu informatycznego, którym dysponuje np. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do systemów informatycznych służb kontrolnych spowoduje, że przepływ informacji będzie szybszy, trafny i bardziej skuteczny, a zarazem tańszy.

Teraz w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej głos zabierze pan poseł Włodzimierz Nykiel.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zmiany kilku aktów prawnych, przede wszystkim ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, bo tego aktu dotyczy prawie 30 zmian, ale także Prawa farmaceutycznego, a ponadto ustaw o drogach publicznych, o transporcie drogowym, o kierujących pojazdami, o Krajowej Administracji Skarbowej, o Policji czy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Celem nowelizacji jest zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów wskazanych w ustawie. Według projektu nastąpi rozszerzenie systemu monitorowania na przewozy kolejowe. W projekcie przewidziano unormowania, które mają łagodzić obowiązek zgłaszania przewozu towaru do odpowiedniego rejestru. Godną odnotowania zmianą wprowadzaną w ramach nowelizacji jest odstąpienie od grupowania towarów zgodnie z polską klasyfikacją towarów i usług. Towary będą oznaczane wyłącznie w oparciu o nomenklaturę scaloną, CN, stosowaną przy wyrobach akcyzowych oraz w obrocie międzynarodowym. Katalog towarów podlegających kontroli rozszerzony został o produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej. Projekt nakłada na przewoźników nowe, obwarowane sankcjami obowiązki, zaś określone organy wyposaża w daleko idące kompetencje. Przepisy nowelizacji przewidują w tym zakresie nowe kompetencje dla generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad. Ważną rolę w projekcie odgrywają przepisy o charakterze sankcyjnym, przewidujące nakładanie kar na podmioty niewywiązujące się z nałożonych obowiązków. Jak było już wskazane w naszym stanowisku podczas pierwszego czytania, sankcje nie tylko mogą dotknąć tych, przeciw którym skierowane są unormowania projektu, tj. podmioty trudniące się nielegalnymi przewozami towarów wrażliwych, ale także mogą dotknąć, i taka jest rzeczywistość, uczciwych przedsiębiorców działających w tej branży, w przypadku których nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków nałożonych ustawą, często szczegółowych i czasochłonnych, powstały np. na skutek przeoczenia. Podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych i Komisji Infrastruktury zwracał na to uwagę także przedstawiciel Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Taki kierunek działań ustawodawcy na pewno zasługuje na aprobatę. Szkoda, że rzadko można się z nim spotkać. Nasz ustawodawca obecnie deklaruje miłość do przedsiębiorcy, ale bardzo chętnie karze go za wiele rzeczy, nakłada sankcje, kary, a także powoduje inne dolegliwości. W toku posiedzenia komisji wiele uwag zgłosili legislatorzy. Podkreślam ich znakomitą pracę. Z drugiej strony oznacza to, że projekt charakteryzował się wieloma wadami w tym zakresie. Biorąc pod uwagę cel regulacji, o której mówię, nasz klub będzie głosował za. Także dodatnio oceniamy pracę komisji. Dziękuję. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! O ile można się zgodzić z założeniami ustawy, że systemy należy uszczelniać, tak jak wskazał pan poseł, o tyle należy brać po uwagę także uczciwych przedsiębiorców, którzy niestety na tej ustawie mogą ucierpieć. Sam projekt nowelizacji ma kilka pozytywnych założeń, ale ma też dwa negatywne. Pierwszym jest wysokość kar sięgających 20 tys. zł, a nawet 100 tys. zł, które mogą dotknąć także przedsiębiorców, którzy mogli nieumyślnie wprowadzić urzędnika w błąd, ale to także kolejne obowiązki dla przedsiębiorców związane z uzupełnianiem zgłoszeń o numery wagonów i pociągów. Natomiast to, co jest najważniejsze w tej ustawie, to to, czego tam brakuje. Brakuje rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców. Jakie to są problemy? Przede wszystkim brak możliwości zgłoszenia korekty zgłoszenia w systemie SENT. Jest to problem, na który zwracają uwagę przedsiębiorcy. Mianowicie w sytuacji popełnienia błędu, ludzkiego błędu, przez człowieka bądź zmiany właściwości zgłoszenia nie ma możliwości dokonania korekty, co może wiązać się z bardzo przykrymi konsekwencjami, nawet wielotysięcznymi karami. Drugą kwestią jest brak wyłączenia stacji paliw spod reżimu ustawy. Ustawa zobowiązuje do zgłaszania przewozu paliw zakupionych przez przedsiębiorcę w chwili zakupu.

Wówczas przedsiębiorca nie ma obowiązku zgłoszenia tego przewozu do systemu SENT, ale jeśli 2 tygodnie później pójdę na tę stację i na podstawie paragonu poproszę o fakturę, a mam takie prawo, wówczas stawiam przedsiębiorcę w niezręcznej sytuacji, bo z jednej strony ma obowiązek - bo ja domagam się faktury - zgłoszenia tego do systemu SENT, z drugiej strony jest już na to za późno, ponieważ on jest zobowiązany do zgłoszenia tego w trybie natychmiastowym. Jeśli chodzi o inny problem, to jest to interpretacja przepisów ustawy. Ustawa bardzo szybko wchodzi w życie, jest bardzo szczegółowa. Kwestia interpretacji. Urzędnicy będą mogli się nauczyć tej ustawy przez 5 lat, bo po 5 latach będą mogli wszczynać kontrolę za 5 lat wstecz z posiadaną wiedzą po 5 latach obowiązywania nowelizacji. Przedsiębiorcy takiego przywileju nie będą posiadali. Na koniec wspomnę też oczywiście o pozytywnych kwestiach. Tą pozytywną kwestią jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów. Pozytywem jest także uproszczenie procedur zgłaszania. Będzie można w ramach jednego zgłoszenia dokonać przewozu różnego rodzaju towarów, jeżeli ten przewóz odbywa się z jednego miejsca do drugiego. Gdy przedsiębiorca naruszy przepisy ustawy, co zostanie ujawnione w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej, kara nie będzie wymierzana, gdy zostanie ustalone, że nie doszło do uszczuplenia należności pieniężnych budżetu państwa. To moim zdaniem jest najważniejsza pozytywna zmiana, dlatego też z uwagi na ten punkt klub Kukiz’15 nie będzie sprzeciwiał się ustawie, będzie rekomendował jej przyjęcie. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, klub Nowoczesna. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Nowoczesna w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw po przedstawieniu sprawozdania komisji. To są druki nr 2156 i 2308. Szanowni Państwo! Przedstawiony Wysokiej Izbie projekt zawiera szereg zmian dotyczących monitorowania przewozu towarów. Co do zasady zmiany te polegają na objęciu monitorowaniem przewozu tzw. towarów wrażliwych realizowanego koleją, odstąpieniu od grupowania towarów zgodnie z polską klasyfikacją wyrobów i usług, pozostaniu przy określeniu rodzaju towarów w oparciu o nomenklaturę scaloną, objęciu systemem monitorowania przewozów produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych określonych w obwieszczeniu, o którym mowa w dotychczas obowiązującym art. 78a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Oczywiście w szczegółach ten projekt był już omawiany podczas zarówno pierwszego czytania, jak i posiedzeń komisji. Te rozwiązania mają swoje ratio legis, w związku z czym większość z nich, powiedziałbym, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno uczciwych przedsiębiorców, jak i strony społecznej i generalnie odpowiada na taką potrzebę pewnego uszczelnienia w tym zakresie. Ale skupię się na tych rzeczach, które są jednak niedobre. Projekt wprowadza również takie rozwiązania właściwie niebezpieczne dla przedsiębiorców, pierwsze, na podstawie którego będzie możliwe wezwanie przewoźnika do przedstawienia środka transportu w określonym miejscu, w określonym czasie, a drugie to absolutnie skandaliczne, drastyczne podwyższenie kar dla uczciwych - i tu pragnę, panie ministrze, jeszcze raz to podkreślić - uczciwych przedsiębiorców branży transportowej. Tu trzeba powiedzieć wyraźnie: rząd PiS chce nakładać kary tylko za to, że przedsiębiorcy nie uzupełnili formularza o jakieś bardzo proste i nieistotne zupełnie dane, jak np. nazwę firmy, a przecież oczywiste jest, że to ma absolutnie drugorzędne znaczenie dla monitorowania przewozów. Tymczasem za brak takiej drugorzędnej informacji rząd PiS chce nakładać nawet 10 tys. zł kary. Gdybyśmy podeszli do tego taktycznie, to należałoby nic nie mówić, tylko poczekać, aż te drakońskie kary zirytują ludzi, natomiast przez ten czas z powodu tego biurokratyczno-finansowego linczu dokonywanego na przedsiębiorcach przez rząd PiS upadłoby wiele polskich firm transportowych.

Miał pan swoje 5 minut, panie pośle. dobro polskich firm transportowych są równie ważne jak dochody budżetowe. Proszę poczytać. Może pan tu przyjść i odpowiedzieć, dlaczego chcecie karać uczciwych przedsiębiorców drakońskimi karami. Jeżeli to jest kłamstwo, to niech pan tu przyjdzie i to powie. Podobne wątpliwości dotyczą sposobu kontroli polegającego na podstawieniu środków transportu na żądanie urzędu. To bardzo istotny temat. Z lektury przepisów można wnioskować, iż jest on całkowicie oderwany od realiów rynkowych i mocno skomplikuje działalność. Otóż należy zauważyć, iż każda firma stosuje swój system organizacji czasu pracy. Wystarczy, że taka informacja dotrze kilka minut po czasie, ktoś jej nie odbierze, ktoś nie przekaże, komuś rozchoruje się dziecko, firma rozładuje towar, po czym otrzyma informację o konieczności podstawienia pojazdu. Być może w związku z tym będzie trzeba zatrudnić nowych pracowników i wzrosną koszty. Zamiast walczyć o rynki Europy nasi przedsiębiorcy walczą z rządem PiS o to, aby w ogóle utrzymać się na rynku. Tu trzeba powiedzieć, że taką postawą państwo absolutnie nie pomagacie naszym firmom w działalności na tych rynkach, gdzie państwa stosują praktyki protekcjonistyczne, i oczywiście na takie postępowanie naszej zgody nie będzie. Warto dobitnie zauważyć, że walka z szarą strefą jest absolutną koniecznością. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wraz z uczciwymi przedsiębiorcami Nowoczesna domaga się właśnie takiej ostrej walki z szarą strefą. Niestety, jak na razie widzimy kolejne obciążenia biurokratyczne i kolejne przeszkody.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Od 18 kwietnia 2017 r. obowiązuje ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Obecny projekt jest poszerzeniem tych zapisów o nadzór nad przewozami kolejowymi i produktami leczniczymi. Oznacza kolejne uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zwiększenie wpływów budżetowych. Jak już dzisiaj zaznaczył pan przewodniczący Komisji Infrastruktury, po zmianach będzie to ustawa o systemie monitorowania przewozów towarów, oczywiście po wprowadzeniu również stosownych zapisów w innych aktach prawnych. Podstawowym celem projektowanej regulacji jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów wrażliwych, takich jak paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym ekodiesel, dodatki do paliw, oleje smarne, odmrażacze na bazie alkoholu, rozcieńczalniki i wiele innych, a także produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.

Kwestia wywozu środków farmaceutycznych i leków to na pewno bardzo istotna sprawa, podnoszona już tutaj w wypowiedziach, jednak tutaj chcę zwrócić uwagę na kwestie związane z tymi zapisami o charakterze restrykcyjnym. To dobrze, że uszczelniamy systemy, że ograniczamy te obszary, mechanizmy i możliwości tam, gdzie przedsiębiorcy stosują różne sposoby, aby obejść konieczność ponoszenia określonych kosztów, jednak tutaj bardzo proszę o rozwagę tak na etapie formułowania myśli i zapisów, jak i później, przy formułowaniu przepisów wykonawczych. W aspekcie całości klub poprze przyjęcie tego projektu. Myślę, że te poprawki, które zostały zgłoszone, czy wątpliwości, które można rozważyć w komisji, będą wyjaśnione.

Panie ministrze, w uzasadnieniu projektu, właściwie w materiałach dołączonych do projektu piszecie państwo o rozwiązaniach stosowanych w innych krajach. Podane są tam przykłady tylko trzech krajów Unii Europejskiej, które zastosowały pewne rozwiązania w odniesieniu do niektórych grup towarów.

Kontrola, monitorowanie dotyczy pewnych tranzytów pewnych tylko rodzajów kawy.

Wysoka Izbo! Nie ulega wątpliwości, że stosowanie tej ustawy jest i powinno być obserwowane, by nie powiedzieć: monitorowane - ale to już w tytule jest monitoring, więc możemy sobie ten termin darować - bo rozszerzenie tego o transport kolejowy było właśnie reakcją na pewne zjawiska. Moje pytanie dotyczy kwestii następującej: Czy stosowanie tej ustawy jest obserwowane i monitorowane od strony ochrony praw przedsiębiorców? Czy obserwując, jak wygląda jej stosowanie, patrzy się także z tego punktu widzenia?

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałem zapytać o restrykcyjność tej ustawy, bo od jakiegoś czasu ta ustawa już funkcjonuje. Tutaj padają dziwne słowa o jakimś linczu na przedsiębiorcach, wręcz o prześladowaniu przedsiębiorców. Czy na skutek działania tej ustawy od jakiegoś czasu, od roku, nastąpiła jakaś upadłość firmy albo czy mają miejsce jakieś dramatyczne sytuacje, które są skutkiem funkcjonowania tej ustawy? Drugie pytanie dotyczy tego procederu zmieniania tras, dziwnych tras.

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jest to oczywiste, że bardzo łatwo jest nakładać kary, bardzo łatwo jest stosować kolejne rozwiązania mające charakter represyjny.

No to ja rozumiem, że chodzi o to, żeby tych przedsiębiorców karać jeszcze bardziej dotkliwie, żeby wpływy do budżetu właśnie z tych kar były jeszcze większe. Jakie, nie wiem, akcje edukacyjne, akcje informacyjne, jakie ich spektrum państwo zastosowali, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, w jaki sposób spełniać te ostre [[Dzwonek]] wymagania? Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan Piotr Walczak. Bardzo proszę.

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Wysoka Izbo! Dziękuję za te pytania, dziękuję również za poparcie tej ustawy. Rzeczywiście de facto ta ustawa funkcjonuje przede wszystkim.

Ale ja zwracam uwagę przede wszystkim na fakt, że. Akurat tak się składa, że w zeszłym tygodniu miałem okazję być w Federacji Rosyjskiej. Rosja także wykazuje zainteresowanie naszymi rozwiązaniami, twierdząc, że są to rozwiązania ciekawe i że rozważy ich wprowadzenie.

Również Litwa zwróciła się do nas o przedstawienie tego systemu.

Zwracam uwagę, że - według tego, co wiem nieoficjalnie - POPiHN nawet chce przyznać Krajowej Administracji Skarbowej tytuł specjalny za wprowadzenie tej ustawy, dlatego że ta ustawa z punktu widzenia przedsiębiorców przede wszystkim powoduje, że są jasne reguły konkurencji. Nie ma przestępców wśród osób handlujących, obracających tymi towarami wrażliwymi.

Podkreślam, że bardzo często zarówno ja, jak i moi współpracownicy spotykaliśmy się z przedstawicielami branży transportu drogowego i branży transportu kolejowego i w ramach tego projektu wypracowywaliśmy właśnie te rozwiązania, które będą korzystne z punktu widzenia nie tylko budżetu państwa, nie tylko wolnej konkurencji, ale także bezpieczeństwa przedsiębiorców. Dlaczego? W związku z tym jeszcze raz chciałem podkreślić, że jak najbardziej jesteśmy w ścisłym kontakcie z przedsiębiorcami, których ta ustawa dotyczy. Bo jeszcze raz chciałem zwrócić uwagę na to, że to nie jest ustawa, która uderza w całą branżę transportową, jeśli w ogóle możemy takiego słowa użyć. To jest ustawa, która dotyczy tak naprawdę niedużej liczby przedsiębiorców, którzy zajmują się przewozem towarów wrażliwych, podkreślam to jeszcze raz: towarów wrażliwych.

Proszę państwa, to jest o tyle ważne, że jako jedyny kraj mamy tak długą granicę lądową z państwami, gdzie papierosy są dużo tańsze.

Ustawa w takiej formie funkcjonuje od ponad roku. Te zmiany, które są, wcale nie powodują zaostrzenia przepisów. To są przede wszystkim rozwiązania, które były postulowane po obserwacji działania tej ustawy przez przedsiębiorców. Co jest najważniejsze? Przez ten rok jej działania nie dotarła do mnie żadna informacja o zniszczeniu polskiego podmiotu, o jakimkolwiek zamknięciu polskiego podmiotu przez Krajową Administrację Skarbową właśnie ze względu na sankcje nałożone przez tę ustawę.

Panie pośle, istnieje tak możliwość, dlatego że istnieje możliwość anulowania starego zgłoszenia i wprowadzenia nowego. Absolutnie nie ma takiej możliwości, że jak ktoś się pomyli w zgłoszeniu, to przedsiębiorca poniesie tego konsekwencje. Jak najbardziej jest procedura, która przez rok funkcjonuje, i nigdy nie było w tym zakresie problemów z jej stosowaniem. Tam są 3 miesiące.

Większość tych rozwiązań funkcjonuje i absolutnie nie jest. Te kwestie, które zauważyliśmy, właśnie w tej ustawie staramy się naprawić. Już w 2017 r. minister finansów wydał w tym zakresie jasną interpretację. Nie ma takich przypadków, takie przypadki się nie zdarzyły. Jest w tym zakresie jasna interpretacja. Dlatego podkreślam - absolutnie i z całą odpowiedzialnością chciałbym to powiedzieć - że nie jest to ustawa, która doprowadziła dzisiaj do jakichkolwiek zaburzeń w branży transportowej, do tego, że jakiekolwiek osoby zbankrutowały.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2290) Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana Michała Wójcika o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę, panie ministrze.

Szanowny Panie Marszałku! Panie Generale! Szanowni Państwo! Mam zaszczyt przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy Kodeks karny wykonawczy, projekt regulacji, które mają usprawnić funkcjonowanie w Polsce systemu dozoru elektronicznego. Tak naprawdę dwa elementy, które są niezwykle istotne, są treścią projektu i na nie chciałbym państwu zwrócić uwagę oraz prosić oczywiście o dalsze prace nad nimi i o ich przyjęcie.

To jest oczywiście również ważne dla osób, które czasami są chronione dzięki temu, że funkcjonuje tenże system. Na podstawie upoważnienia ustawowego minister sprawiedliwości będzie miał możliwość zdecydować, że Służba Więzienna będzie mogła być podmiotem, który nie tylko obsługuje centralę monitorowania skazanych. Dzisiaj takie zadanie ona wykonuje.

Tak jest dzisiaj, kiedy wykonuje te zadania konsorcjum na podstawie podpisanej umowy. Oczywiście otrzymuje ono określone środki, wykonując te zadania. Są tzw. patrole kontrolujące funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, no i czasami oczywiście trzeba działać. Problem polega tylko na tym, że podmiot prywatny nie dysponuje takimi uprawnieniami, żeby np. zatrzymać daną osobę, tylko zazwyczaj musi wzywać policję. Tu jest istotna słabość całego systemu. A Służba Więzienna, funkcjonariusze Służby Więziennej mają oczywiście prawo stosować różnego rodzaju środki przymusu bezpośredniego. Oczywiście kwestią fundamentalną jest to, jaką filozofię mamy, jeżeli chodzi o sprawę związaną z funkcjonowaniem tego rodzaju systemu.

Po drugie, ten system musi być również korzystny z punktu widzenia gospodarczego.

Jeżeli chodzi o kwestię drugą, czyli usprawnienie tego całego systemu, to chodzi o zastosowanie tzw. rejestratora przenośnego.

Ona musi mieć rejestrator, tak jak w przypadku systemu stacjonarnego, gdzie jest rejestrator, gdzie w sytuacji, kiedy widzimy, że coś się dzieje, że osoba np. łamie zakaz. Zazwyczaj to jest tak, że jakaś odległość w metrach jest przewidziana, ta osoba musi się poruszać, zazwyczaj to jest w postanowieniu określone, w jakich dniach tygodnia, w jakich godzinach.

A jeżeli mamy system dozorujący o charakterze zbliżeniowym, mobilnym, to tutaj już tych rejestratorów nie mamy, czyli jedyny sygnał, który możemy dać. Dochodzi do wibracji dających sygnał, że coś się dzieje, że coś jest naruszane, jakiś zakaz, ale nie możemy się skontaktować z daną osobą. Dlatego chcemy, żeby taki rejestrator te osoby posiadały, żeby ten system był już kompletny, czyli żeby można było się łączyć, wydawać polecenia za pomocą rejestratora przenośnego, żeby ta osoba tym rejestratorem dysponowała.

Chcemy także znowelizować jeden z przepisów, rozszerzając de lege ferenda zakres zastosowania dozoru elektronicznego również na środki inne niż środki karne i środki zabezpieczające. Chodzi o rozszerzenie funkcjonalności systemu dozoru elektronicznego w przyszłości, nie możemy wykluczyć, że będą zmiany w tym zakresie również podejmowane, a więc już taki przepis jak najbardziej pojemny twórzmy, żeby rzeczywiście ten system działał. Muszę powiedzieć, że jeżdżę na różne spotkania, spotykam się z ludźmi, oni często pytają: Panie ministrze, jak to jest z tym systemem dozoru elektronicznego, dlaczego nie rozpowszechniać go? Oczywiście, że staramy się go upowszechniać w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze skazanymi. Pamiętajmy, że było w ogóle załamanie, jeżeli chodzi o stosowanie tego systemu, jest kwestia stosowania go, tylko jeżeli chodzi o karę ograniczenia wolności. My wróciliśmy w czasach dobrej zmiany do tego, żeby go stosować, jeżeli chodzi o kary pozbawienia wolności. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ten system był jak najbardziej rozszerzany, bo nie chodzi nam o to, żeby wypełniać ludźmi więzienia. Dlaczego? Lepiej jest, jeżeli człowiek np. w ramach systemu dozoru elektronicznego wykonuje w warunkach wolnościowych karę pozbawienia wolności, bo może pracować.

Oczywiście prowadzimy także prace analityczne w ministerstwie, jeżeli chodzi o kwestię rozszerzenia katalogu osób, co do których można by było zastosować system dozoru elektronicznego. Natomiast ta zmiana jest zmianą fundamentalną, bo ona pokazuje, że dzisiaj inaczej będziemy patrzyli na cały system. Oczywiście mieszany może być, bo przepis daje takie prawo, to jest ta furtka, że w przyszłości jeżeli ktoś zastosuje przepisy zamówień publicznych, będzie miał taką możliwość, żeby wybrać podmiot prywatny. Ale co do zasady dajemy szansę, żeby również to wykonywał podmiot o charakterze czysto publicznym - w tym przypadku chodzi o Służbę Więzienną. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Bartłomiej Wróblewski.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy Kodeks karny wykonawczy, druk nr 2290. Zgadzamy się z celami, które przyświecały Radzie Ministrów przy przygotowaniu tego projektu. Są nimi zwiększenie kompetencji Służby Więziennej w ramach systemu dozoru elektronicznego, a także poszerzenie w tym systemie możliwości wykorzystania rejestratorów przenośnych. Skutkiem nowelizacji będzie ustawowe umocowanie ministra sprawiedliwości do fakultatywnego powierzania wykonania zadań, o których mowa w art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego, właśnie Służbie Więziennej. Uważamy, że zagwarantuje to nieprzerwane i sprawne wykonywanie kar w systemie dozoru elektronicznego. W przypadku decyzji ministra sprawiedliwości Służba Więzienna przejmie od podmiotu komercyjnego całość zadań podmiotu dozorującego, które obejmują wykonywanie całodobowych patroli interwencyjnych przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej na terenie całego kraju z zabezpieczeniem przez Służbę Więzienną niezbędnych środków transportu i łączności oraz bezpiecznego transferu danych między zespołami patrolowymi a Centralą Monitorowania Systemu Dozoru Elektronicznego, związanych z wykonywaniem kar, środków karnych i zabezpieczających. W efekcie nawet w przypadku wystąpienia poważnych zdarzeń krytycznych, kiedy to upoważniony podmiot dozorujący zaprzestanie wykonywania kar w SDE, nowa regulacja umożliwi sprawne i pilne przejęcie ich realizacji przez Służbę Więzienną. To jest kluczowy argument w tej sprawie. Także w przypadku modyfikacji funkcjonowania SDE w przyszłości proponowana regulacja pozwoli na elastyczniejsze zarządzanie tym systemem.

Zaopatrzenie skazanego w rejestrator przenośny nie tylko umożliwi kontakt telefoniczny z organami dozorującymi, ale też zapewni kontrolę jego miejsca pobytu w czasie rzeczywistym nawet w przypadku wyczerpania się źródła zasilania w podstawowym urządzeniu telefonicznym, jakim jest obecnie nadajnik GPS.

Ta sprawa musi być wprost uregulowana w ustawie.

Pan poseł Michał Szczerba, klub Platforma Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! System dozoru elektronicznego pozwala na stałe i dyskretne kontrolowanie zachowania osoby skazanej. Sąd wyznacza jej obowiązki. Zgodnie z podanym harmonogramem osoba poddana kontroli musi np. przebywać w domu lub w innym miejscu odbywania kary w ściśle określonych godzinach. Szanowni Państwo! Dotychczas Służba Więzienna wykonywała pewne zadania ustawowe związane z odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego. Dotyczyły one głównie prowadzenia centrali monitorowania. Zdaniem rządu kompetencje Służby Więziennej powinny zostać poszerzone również o prawo do realizacji innych zadań immanentnie związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że wykorzystywanie rejestratorów przenośnych w ramach systemu dozoru elektronicznego jest w Polsce niewielkie.

Mogłoby być tego o wiele, wiele więcej. Chciałbym zwrócić uwagę, że jest to system bardzo korzystny. Przede wszystkim umożliwia on skazanym zachowanie więzi z rodziną, wykonywanie pracy zarobkowej, zmniejsza też zaludnienie jednostek penitencjarnych.

Brak istnienia, tak naprawdę, efektywnej służby zdrowia. Były liczne zaniedbania proceduralne, których najlepszym przykładem w tej kadencji była sprawa pani Agnieszki Pysz, która zmarła w areszcie śledczym na Grochowie, kiedy nie udzielono jej skutecznej pomocy medycznej, ignorowano jej błagania o jej udzielenie. Następnie tę sprawę skierowano do wyjaśnienia kierownikowi ambulatorium, który nie podejmował tego skutecznego leczenia. To są wielkie zaniedbania, dlatego też system dozoru elektronicznego jest również pewnym ważnym wyzwaniem. Druga sprawa to są wystąpienia, które kierują w sprawie dozoru elektronicznego zarówno rzecznik praw obywatelskich, jak i rzecznik praw dziecka. To są wystąpienia, które dotyczą przede wszystkim częstszego wykorzystania tego systemu w sprawie przestępstwa niealimentacji.

Jak powiedziałem, jest to decyzja rządu, aby tego dozoru nie wykonywał podmiot dozorujący, czyli podmiot zewnętrzny, jak było dotychczas. Intencją rządu jest to, żeby te działania wykonywała sama Służba Więzienna. My przyjmujemy to stanowisko jako informację, a o naszym podejściu do sprawy poinformujemy Wysoki Sejm w terminie późniejszym. Pani poseł Barbara Chrobak, klub Kukiz’15. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Nieudolne działanie Platformy Obywatelskiej doprowadziło w 2015 r. do drastycznego spadku orzeczeń o wykonywaniu kary w SDE i w rezultacie do zmarginalizowania tej instytucji w sferze polityki karnej. Dozór elektroniczny stał się za sprawą reformatorów z PO rodzajem kary ograniczenia wolności, a nie jak wcześniej sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności. Szczerze powiedziawszy, wzbudziło to nasze zdziwienie, bo było to chyba jedyne działanie PO i PSL wymierzone przeciwko przestępcom, oczywiście nie tym groźnym, ale tym najdrobniejszym: niepłacącym alimentów, kierującym pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości, sprawcom przestępstw zniszczenia mienia i gróźb karalnych. O tych grubych graczy wyłudzających podatki, organizujących lunaparki VAT-owskie, przedsiębiorców hazardowych i Platforma nigdy nie zapomniała zadbać. Było to w rezultacie działanie wymierzone przeciwko interesom ekonomicznym państwa, bo spadek liczby orzeczeń o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w SDE skutkował wzrostem kosztów utrzymania więźniów w zakładach karnych. Krótko mówiąc, Platforma Obywatelska razem z PSL-em wolała wydawać 3,5 tys. zł na utrzymanie więźnia niż 330 zł na koszty utrzymania skazanego poza jednostką penitencjarną w SDE. Obecny rząd, i słusznie, dokonał zmiany przepisów i powrotu do rozwiązań sprzed 1 lipca 2015 r. W rezultacie wzrosła ilość kar pozbawienia wolności wykonywanych w SDE. Utrzymywanie skazanych za drobne przestępstwa w zakładach karnych jest bowiem nieopłacalne nie tylko ekonomicznie, ale i społecznie. Nie jest tajemnicą, że izolacja w warunkach zakładu karnego z kryminologicznego punktu widzenia niczego dobrego nie uczy, wręcz przeciwnie, stygmatyzuje, wyrywa z więzi społecznych, powoduje utratę pracy, a często rozpad rodziny. Sprawne wykonywanie kar w SDE wymaga jednak stałego monitoringu, także niezbędnych korekt legislacyjnych. W tym kierunku zmierza nowelizacja. Nie budzi wątpliwości klubu Kukiz’15 szerokie powierzenie Służbie Więziennej dotychczasowych wyłącznych kompetencji ministra sprawiedliwości w zakresie wykonywania zadań związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności w SDE. Dotychczas, szanowni państwo, funkcjonujący system uniemożliwiał kontakt ze skazanym w dozorze mobilnym za pośrednictwem urządzenia zainstalowanego na kończynie. Obecnie proponuje się wyposażenie skazanego w rejestrator przenośny umożliwiający taki kontakt, co w konsekwencji zapewni zwiększoną kontrolę w trakcie wykonywania kary w SDE. Oczywiście takie techniczne rozwiązanie wymaga dodatkowej obudowy prawnej, a w szczególności usankcjonowania prawnego obowiązku po stronie skazanego do odbierania połączeń. Pracując przez wiele lat w wymiarze sprawiedliwości, spotykałam się często z problemami wynikającymi ze stosowania wolnościowych środków zapobiegawczych. Najlepszym przykładem wydaje się tu dozór Policji. W bardzo wielu przypadkach środek ten okazywał się fikcyjny, podobnie jak zobowiązanie podejrzanego do przebywania w określonym miejscu czy zakaz opuszczania kraju. Podejrzani często nie wykonywali ani nie wykonują tych obowiązków. Prokuratorzy nadzorujący postępowania przygotowawcze dowiadywali się o tym z dużym opóźnieniem. Stanowi to nierzadko istotne zagrożenia dla podstawowej przesłanki stosowania środków zapobiegawczych, jaką jest zabezpieczenie prawidłowego toku prowadzenia postępowania. Stąd też de lege ferenda - takie prace, jak wiadomo, trwają - za niezbędne uznać należy objęcie systemem dozoru elektronicznego wolnościowych środków zapobiegawczych. Taki monitoring zapewni natychmiastowy przekaz, że np. podejrzany nie stawia się na dozór, a w dalszej konsekwencji reakcję prokuratora nadzorującego postępowanie, który będzie mógł w celu zabezpieczenia jego prawidłowego toku rozważyć zatrzymanie i zastosowanie surowszych środków, włącznie z tymczasowym aresztowaniem. Reasumując, panie marszałku, Wysoka Izbo, widać po tym projekcie, że w odróżnieniu od państwa z Platformy Obywatelskiej, która, o dziwo, tym razem nie zadbała o swój popadający w konflikt z prawem elektorat, obecne kierownictwo resortu sprawiedliwości interesuje się SDE, unowocześnia go oraz zwiększa jego funkcjonalność techniczną i prawną. Pan poseł Mirosław Suchoń, klub Nowoczesna. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Nowoczesna w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy Kodeks karny wykonawczy, zawartego w druku nr 2290. Szanowni Państwo! Projekt dotyczy de facto dwóch obszarów funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego. W pierwszym zakresie przedstawiony przez rząd projekt ma na celu szerokie umożliwienie Służbie Więziennej wykonywania zadań związanych z odbywaniem kary właśnie w systemie dozoru elektronicznego.

Natomiast w projekcie rząd proponuje poszerzenie kompetencji Służby Więziennej o inne zadania, kompleksowo zdefiniowane w art. 43t Kodeksu karnego wykonawczego. Miałoby to polegać na ustawowym umocowaniu ministra sprawiedliwości w zakresie fakultatywnego powierzania wykonywania zadań podległej sobie Służbie Więziennej. Co oczywiste i co jest konsekwencją takiego projektu, scedowanie przez ministra sprawiedliwości zadań podmiotu dozorującego na Służbę Więzienną nie odbywałoby się w ramach Prawa zamówień publicznych. Oczywiście, jak pan minister wspomniał w trakcie prezentacji tego projektu, jest to pochodna innej wizji systemu dozoru elektronicznego, ponieważ do tej pory część tych zadań wykonują firmy, natomiast z tego, jak należy rozumieć ten projekt i co przedstawił pan minister, wynika, że rząd zmierza do powierzenia wszystkich czynności wyłącznie jednostkom, które będą jednostkami publicznymi, takimi jak właśnie Służba Więzienna.

Te przepisy również są zawarte w projekcie, i to dobrze.

Tu jest zawsze takie niebezpieczeństwo, panie ministrze, że może zostać to użyte w bliżej nieokreślonym celu, dlatego Nowoczesna wnosi o skierowanie tego projektu do dalszych prac w komisji, natomiast w trakcie tych prac będziemy prosić o to, żeby dokładnie wytłumaczono, z czym te przyszłościowe zadania mogą się wiązać, tak żeby mieć również na uwadze prawa obywatelskie, które w ramach tych przepisów muszą być przestrzegane. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Panie Generale! Wysoka Izbo! Przygotowana nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej w swym założeniu ma na celu szerokie umożliwienie tej formacji wykonywania zadań związanych z odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego. Służba Więzienna w chwili obecnej wykonuje jedynie zadania ustawowe, wskazane przez ministra sprawiedliwości, które sprowadzają się jedynie do prowadzenia centrali monitorowania w SDE. Jak wynika z wieloletniej praktyki funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego, ma on charakter bardzo ograniczony, a zatem wymaga to poszerzenia kompetencji Służby Więziennej również o prawo do realizacji innych zadań immamentnie związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności w systemie dozoru elektrycznego. Dotychczas zadania te zostały kompleksowo zdefiniowane przez ustawodawcę w Kodeksie karnym wykonawczym, czego dowodzi zapis art. 43t. Wskazuje on zadania możliwe do realizacji wyłącznie przez upoważniony podmiot dozorujący. Przedłożony projekt ustawy zakłada zmianę tego stanu rzeczy poprzez ustawowe umocowanie ministra sprawiedliwości do fakultatywnego powierzania wykonywania zadań, o których mowa we wspomnianym powyżej przepisie Kodeksu karnego wykonawczego, podległej sobie formacji mundurowej, jaką jest Służba Więzienna. Jak przekonuje resort sprawiedliwości, ma to zagwarantować pełną spójność w zakresie nieprzerwanego oraz sprawnego wykonywania orzeczonych kar w systemie dozoru elektronicznego, i to nawet w sytuacjach poważnych zdarzeń krytycznych, kiedy to upoważniony podmiot dozorujący, np. prywatny, zaprzestanie wykonywania rzeczonych kar w SDE. Nowa regulacja ustawowa miałaby w takich przypadkach umożliwić sprawne i pilne przejęcie realizacji dotychczasowych zadań tego podmiotu przez Służbę Więzienną. Projektodawcy ustawy przewidują, iż w przypadku modyfikacji funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w przyszłości, przewidzianej nowelizacją przepisu art. 43a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego np. o poszerzenie zakresu stosowania SDE o środki zapobiegawcze, proponowana regulacja pozwoliłaby na elastyczne zarządzanie tym systemem. Zamierzony cel mógłby zostać niezwłocznie osiągnięty, albowiem już bez wymogu dodatkowych uzgodnień, aneksowania oraz uzgadniania nowych zapisów umownych zadania te byłby przejęte i realizowane właśnie przez Służbę Więzienną. Resort proponuje uchylenie oraz znowelizowanie kilku zapisów ustawy o Służbie Więziennej i jednocześnie podkreśla zasadność umocowania ministra sprawiedliwości właśnie do fakultatywnego powierzania wykonywania zadań formacji mu podległej lub przez niego nadzorowanej. Nowelizacja zakłada także zmianę przepisu związaną z poprawą funkcjonalności urządzeń związanych z dozorem mobilnym. Jak wskazuje resort, do tej pory skazany w dozorze mobilnym wyposażony był jedynie w nadajnik GPS, montowany na kończynie, który z uwagi na swoją konstrukcję techniczną nie pozwalał na nawiązanie kontaktu telefonicznego pomiędzy organami dozorującymi a skazanym. Wyposażenie zatem skazanego w rejestrator przenośny umożliwi mu taki kontakt, a także pozwoli na kontrolę miejsca pobytu skazanego w czasie rzeczywistym, nawet w przypadku wyczerpania się źródła zasilania w nadajniku GPS. W przekonaniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów każda zmiana służąca dobru państwa lub jednostki zasługuje na poparcie, jednakże zakres przedmiotowy i cele tej regulacji winny zostać bardzo szczegółowo, z najwyższą ostrożnością, dogłębnie przeanalizowane, i to po zasięgnięciu opinii zarówno Sądu Najwyższego, jak i generalnego inspektora ochrony danych osobowych, tak aby pracując w niezwykłym pośpiechu, ustrzec się błędów, które często są nie do naprawienia. Analizy i wyjaśnienia wymaga także sytuacja wpływu ewentualnego uchwalenia projektu na działalność gospodarczą, stąd opowiadamy się za skierowaniem projektu ustawy do dalszych prac parlamentarnych. Do zadania pytań zgłosiło się pięcioro pań i panów posłów. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Paweł Bańkowski, klub Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zgodnie z treścią uzasadnienia projektowanej ustawy w przypadku powierzania zadań podmiotu dozorującego bez zastosowania Prawo zamówień publicznych jednostce organizacyjnej podległej ministrowi sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej innej niż Służba Więzienna jednostka taka będzie spełniać przesłanki udzielenia zamówienia in-house. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych tzw. zamówienia in-house są zamówieniami udzielanymi w trybie zamówienia z wolnej ręki, który nie stanowi o wyłączeniu stosowania Prawo zamówień publicznych, a jedynie przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z jedynym wykonawcą w celu udzielenia zamówienia. I pytanie, panie ministrze: Co w takim przypadku autorzy projektowanej ustawy przewidują, jaka będzie realność prowadzenia negocjacji pomiędzy ministrem sprawiedliwości a podległą mu służbowo lub nadzorowaną przez niego jednostką organizacyjną w celu udzielenia przedmiotowego zamówienia, mając na uwadze zwłaszcza zasadę racjonalnego wydatkowania środków publicznych? Pytanie zadaje pani poseł Małgorzata Pępek, Platforma Obywatelska. Panie Ministrze! Chodzi o wyposażenie skazanego na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego w rejestrator przenośny. Ma to pozwolić na kontrolę miejsca pobytu skazanego w czasie rzeczywistym, nawet w przypadku wyczerpania się baterii nadajnika. Projekt, jak czytamy w uzasadnieniu, powoduje skutki dla budżetu państwa.

Pytanie zadaje pan poseł Jerzy Meysztowicz, klub Nowoczesna. Bezpośrednio z ustawy to nie wynika, ale z wypowiedzi pana ministra wynika, że tak na dobrą sprawę cały system będzie docelowo przekazany Służbie Więziennej. Ja nie uważam, żeby to było złe rozwiązanie.

Czy dochodziło do jakichś nieprawidłowości i to było powodem, dla którego państwo zdecydowaliście się na to, że cały ten system zostanie włączony w działania Służby Więziennej? Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pani poseł Zofia Czernow, klub Platformy Obywatelskiej. Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Po pierwsze, czy ten projekt ustawy oznacza, bo nie jestem tego pewna, że Służba Więzienna będzie jedynym nadzorującym odbywanie kary w SDE, czy też będą możliwe mieszane formy odbywania kary? To pierwsze pytanie.

Bardzo dziękuję.

Na jakie straty będą narażone te firmy, jeżeli całość obsługi zostanie przejęta przez Służbę Więzienną?

W związku z tym jakie państwo poczyniliście kroki, żeby ten system był sprawniej wykorzystywany, czy w ogóle jakieś kroki zostały poczynione? Wysoki Sejmie! Na galerii witamy młodzież z powiatu rawskiego. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Głos zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pan Michał Wójcik.

Szanowny Panie Marszałku!

Dziękuję bardzo za włączenie się w dyskusję. Najpierw odpowiem panu posłowi Bańkowskiemu.

Po prostu minister sprawiedliwości poleci podległej służbie, w tym przypadku Służbie Więziennej, wykonywanie tych zadań i te zadania będą wykonywane, tu nie wchodzi w grę żaden przepis ustawy o zamówieniach publicznych.

Dlaczego? Firma z jakichś powodów, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, może odstąpić od wykonania umowy, a przecież pamiętajmy, jakie zadanie jest realizowane. W tle mamy nadzór nad osobami, które weszły w kolizję z prawem.

To jest bardzo dobre pytanie.

Natomiast jest jedna rzecz, która jest istotna, szanowni państwo. Zgodnie z ustawą są określone warunki, kiedy można stosować ten system. Jest kategoria podmiotów, które mogą wystąpić o to, żeby zastosować dozór elektroniczny, to raz. Trzy, cele kary muszą być zrealizowane, bo to jest bardzo istotna sprawa.

Czy nie będzie strat dla firm? Jeszcze raz mówię, że jeżeli chodzi o wykonanie tego zadania w ramach podpisanej umowy, to będzie ono realizowane do końca września 2018 r. Jeżeli decyzja zostanie podjęta, oczywiście jeżeli chodzi o wykonywanie tego zadania przez Służbę Więzienną, zadanie to będzie realizowane - rozumiem, że panu posłowi chodziło o to, że wówczas firma komercyjna nie będzie tego wykonywała.

To jest kwestia dotycząca zdarzenia, które miało miejsce w jednym z zakładów karnych. Chcę państwu powiedzieć, że zostały wyciągnięte bardzo daleko idące konsekwencje wobec dyrektora tego zakładu karnego w Warszawie.

Sprawa druga to jest kwestia tego zaplecza medycznego w Służbie Więziennej.

Na służbę medyczną - to zabezpieczenie, o którym mówił pan poseł Szczerba - nigdy w historii nie wydano takich pieniędzy, jak w ostatnim czasie.

Ci, którzy są lekarzami, świetnie o tym wiedzą. Chcę powiedzieć, że bardzo duże pieniądze poszły na służbę medyczną w ramach zakładów karnych. Nigdy takich modernizacji nie było. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście stan polskiego więziennictwa, więzień, infrastruktury jest fatalny. On był zaniedbywany przez dziesiątki lat.

Jeżeli chodzi o kwestie. Ach, ważne jest pytanie, które padło ze strony chyba pana posła Bańkowskiego albo pana posła Suchonia, już nie pamiętam dokładnie, przepraszam bardzo, o kwestię środków zapobiegawczych, czyli o stworzenie przepisu na przyszłość.

O co chodzi? Chodzi o to, żeby ewentualnie można było zastosować ten system do innych środków zapobiegawczych, np. dozoru policyjnego, tymczasowego aresztowania. Dzisiaj jeszcze ustawodawca nad tym nie pracuje, ale to nie zabrania nam przecież pracy w tym zakresie. I to nie jest błędne od strony legislacyjnej. To jest, wydaje mi się, wszystko.

Nam nie chodzi o to, i my to bardzo mocno podkreślaliśmy, zmieniając art. 209 Kodeksu karnego, czyli tam, gdzie wyłączyliśmy przesłanki uporczywości, jeżeli chodzi o niezaspokajanie podstawowych potrzeb osoby uprawnionej, podstawowych potrzeb życiowych. Wiemy o tym doskonale. Chodzi o to, żeby oni pracowali i żeby mogli rzeczywiście zaspokajać te podstawowe potrzeby.

Dzisiaj już się tak prosto nas nie oszuka, że ktoś nie ma pracy i po prostu nie ma możliwości podjęcia działań zarobkowych, żeby wywiązać się np. w stosunku do osoby uprawnionej. Tak że prosiłbym bardzo serdecznie Wysoką Izbę o dalsze prace nad tym projektem. Będziemy starali się szczegółowo informować państwa o tym, co się kryje pod każdym z proponowanych przepisów.

Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy Kodeks karny wykonawczy, zawarty w druku nr 2290, do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 1607 i 1928) Proszę panią poseł Iwonę Śledzińską-Katarasińską o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Rozwiązania zawarte w druku nr 1928, oparte na senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, dotykają bardzo ważkiego społecznie problemu i są dowodem próby zmniejszenia nierówności, zlikwidowania barier dla osób, które z przyczyn całkowicie od siebie niezależnych nie mogą w pełni korzystać z bogactwa życia codziennego.

Ta sprawa jest znana od lat. Oczekiwania tych środowisk są w pełni uzasadnione, słuszne. Przypomnę, że w tej chwili rozwiązanie prawne zobowiązuje nadawców programów telewizyjnych do zagwarantowania 10% czasu w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyjątkiem oczywiście reklam i telesprzedaży, w taki sposób, by te osoby, o których tutaj mówimy, mogły z tego programu korzystać. Oczywiście 10% to jest coś, ale trudno powiedzieć, czy to jest kres oczekiwań czy aspiracji tego środowiska, które ma prawo w pełni uczestniczyć, tak jak osoby, które słyszą dobrze, widzą dobrze, w życiu kulturalnym, a telewizja w jakimś sensie jest także wyznacznikiem życia kulturalnego.

Komisja pracowała w ścisłym kontakcie i powiązaniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz ministerstwem kultury, bo w gruncie rzeczy ta ustawa - mam nadzieję, że będzie przyjęta przez Wysoką Izbę - nakreśla tylko pewne ramy, a tak naprawdę jej realizacja będzie zależała od rozporządzenia, jakie przedstawi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Tak było do tej pory, tak jest i tak będzie w przyszłości. O wadze tego tematu i o tym, że staraliśmy się - mimo że, jak mówię, otrzymaliśmy projekt z Senatu - jako komisja bardzo poważnie podejść do tej kwestii, świadczy choćby to, że została powołana podkomisja.

To oczywiście było ciągle za mało, ale tak jak mówię, uznaliśmy, że w tej chwili w perspektywie najbliższych 5 lat jest to kres możliwości, aczkolwiek - może nie wypada zaczynać sprawozdania od końca - chcę zwrócić uwagę na art. 4, który wprowadziła komisja, to jest rozwiązanie, którego w ogóle nie było w projekcie senackim, który stanowi, że w roku 2025 przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przedstawi Sejmowi, Senatowi oraz ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o realizacji obowiązków, które są określone w tym projekcie, a także możliwości zwiększenia poziomu udogodnień w programach telewizyjnych. Myślę, że ten art. 4, aczkolwiek można powiedzieć, że jest w jakimś sensie deklaratywny, pokazuje, że zarysowany w projekcie ustawy poziom 50-procentowego udziału programów z wszelkiego rodzaju udogodnieniami nie jest poziomem granicznym.

Wraz z rozwojem techniki będzie możliwe znaczne podwyższenie tego poziomu.

A więc to są elementy dźwiękowe lub graficzne, które dają możliwość zapoznania się z audycją, w szczególności w formie napisów dla niesłyszących lub audiodeskrypcji, a także tłumaczenia na język migowy.

Ze swej strony mogę tylko powiedzieć, że dla mnie właściwa praca nad realizacją tej ustawy zacznie się na etapie konsultacji, pewnego rodzaju negocjacji środowisk osób niesłyszących, niewidzących, niedosłyszących, niedowidzących z krajową radą, bo to jest problem, ile czego. Jak wiadomo, pewne formy są tańsze dla nadawcy, inne są droższe, w bezpośrednim przekazie o pewne formy jest łatwiej, o inne formy jest trudniej, a tak jak mówię, te formy to albo audiodeskrypcja, albo język migowy, albo napisy. Art. 2 - tutaj w stosunku do rozwiązań proponowanych przez Senat musieliśmy wprowadzić pewne zmiany, ponieważ przesunęło się w czasie.

Musieliśmy zmienić kalendarium. Ono jest zmienione, ale też rozpisane niejako na lata.

Ta zmiana w kalendarium sprawiła, że musieliśmy jeszcze raz przemyśleć, kiedy wchodzą w życie poszczególne przepisy, a kiedy tracą moc dotychczasowe.

Pewne przepisy tracą moc 31 marca 2019 r., a ustawa sama w sobie wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, przy czym oczywiście te przepisy z rozporządzenia, które są obwarowane karami dla nadawców, mogą wejść w życie dopiero 1 stycznia 2019 r. To daje krajowej radzie możliwość przystąpienia wcześniej do prac studyjnych i negocjacji, przygotowania tych rozporządzeń, tak żeby potem, 1 stycznia, to wszystko zaskoczyło.

On pozornie wygląda niezbyt okazale, ale myślę, że jest projektem, nad którym warto było tak szczegółowo się pochylić. Chciałam, korzystając z okazji, podziękować wszystkim, którzy wspomagali zarówno podkomisję, jak i komisję w szukaniu tych najlepszych, najbardziej precyzyjnych rozwiązań.

To prawda, ale przyznaję szczerze, że tu polegliśmy i tego słowa „udogodnienia” nie umieliśmy niczym innym równie precyzyjnym z punktu widzenia prawnego i legislacyjnego zastąpić.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Serdecznie państwa pozdrawiamy. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Bardzo proszę, panie pośle. Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Wysoka Izbo! Miarą rozwoju cywilizacyjnego państwa jest m.in. stosunek do niepełnosprawnych. Elementem integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem jest dostęp do informacji, do mediów. Szczególnie dotyczy to ludzi z dysfunkcjami wzroku, słuchu. Tych pierwszych jest w Polsce ok. 300 tys., tych drugich - ok. 100 tys., a więc niemała grupa, i dla nich telewizja jest ważnym źródłem informacji. Jak słyszeliśmy dzisiaj, ustawa mówi o 10% programów z udogodnieniami dla niepełnosprawnych. Na szczęście realnie jest znacznie lepiej. Na przykład według informacji telewizji publicznej w pierwszym programie już ok. 50% emisji to emisje z udogodnieniami, w drugim programie - ok. 30%, a na kanale TVP Seriale - nawet 80%. Zresztą w telewizjach komercyjnych też jest to procent znacznie wyższy niż te ustawowe 10%. Oczywiście dosyć daleko nam jeszcze do najbardziej rozwiniętych krajów, które, po pierwsze, są bogatsze, a po drugie, już lata temu zaczęły prowadzić intensywne prace nad udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Ta ustawa jest pokłosiem petycji, która trafiła do Sejmu do komisji petycji.

Te dyskusje pokazały, że rzecz jest na tyle skomplikowana, że sejmowa komisja petycji nie jest w stanie podołać technicznie, organizacyjnie, merytorycznie temu zadaniu. Natomiast na szczęście na podstawie jednobrzmiącej petycji z inicjatywą ustawodawczą zdecydował się wystąpić Senat. Projekt był bardzo szeroko konsultowany przez różne środowiska, omawiany w komisji, w podkomisji nadzwyczajnej.

To są w skali roku wielomilionowe koszty na jedno tylko pasmo.

Szczególnie liczę tutaj na rozwój technologiczny, rozwój techniczny, który dzięki nowym urządzeniom [[Dzwonek]] pozwoli ten procent udogodnień zwiększyć.

Bardzo proszę, pani poseł Elżbieta Gapińska, Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo!

Musieliśmy podjąć pewne działania związane z tym, żeby rzeczywiście dobra kultury, tak jak już tutaj mówiła przewodnicząca podkomisji, pani poseł Śledzińska-Katarasińska, zostały udostępnione tym osobom w większym zakresie, niż to miało miejsce dotychczas, bo dotychczas, jak państwo doskonale wiecie, było to tylko 10%, które było wymagane, 10%. W tej chwili podjęliśmy decyzję, żeby docelowo te udogodnienia miały miejsce na poziomie co najmniej 50%, ale „co najmniej” nie oznacza, że jest to granica górna.

Mówię to szczególnie do tych osób, które są niepełnosprawne i które zwracały się do nas w mailach, w pismach, mówiły o tym, że to jest niewystarczające udogodnienie. Oczywiście będzie to przejrzane przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który w roku 2025 ma złożyć sprawozdanie na ręce senatorów, posłów oraz ministerstwa, w jaki sposób ta ustawa jest realizowana przez media.

Myślę, że to jest możliwe do osiągnięcia, a być może nawet stanie się to wcześniej. Może właśnie będzie tak ze względu na możliwości techniczne, więc miejmy taką nadzieję. Na pewno jesteśmy tutaj zdecydowani, tak jak pracowaliśmy w konsensusie w podkomisji, gdzie właściwie wszyscy przedstawiciele podkomisji niezależnie od tego, z jakich środowisk się wywodzili, byli zdecydowani, żeby takie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami uchwalić. Dlatego pełna dobrych nadziei na to, że być może nawet szybciej niż w tym roku 2024 uda się osiągnąć ten poziom 50%, w imieniu klubu Platforma Obywatelska chcę zadeklarować, że nasz klub będzie oczywiście popierał ten projekt i będziemy za nim głosować, bo uważamy, że jest niezwykle potrzebny. Bardzo proszę, pani poseł Elżbieta Zielińska, klub Kukiz’15. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus, klub Nowoczesna. W zasadzie cóż tutaj można więcej dodać po wypowiedzi mojej koleżanki? My wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że ten projekt powinien powstać już wcześniej, że to powinno już się wydarzyć, a żadna z osób, szczególnie osoby głuche, słabo słyszące, niewidome, nie powinna być dyskryminowana. Mówimy o 4 mln dyskryminowanych obywateli i powinniśmy zrobić wszystko, aby nie tylko ta ustawa weszła w życie jak najszybciej, nawet zakładając, że te zmiany będą postępowały w ciągu następnych kilku lat. Pomimo wszystko powinniśmy zrobić tak, aby jednak przyspieszyć te prace ze względu właśnie na to, że mamy do czynienia z tak dużą liczbą obywateli. My jako klub Nowoczesna oczywiście będziemy głosowali za tym projektem, ale też jako klub Nowoczesna będziemy domagali się tego, aby jednak przyspieszyć prace nad wdrożeniem dostępności telewizji szybciej, niż to teraz zakładamy. W zasadzie mogę tutaj obiecać naszą pomoc przy pracach i mam nadzieję, że będzie taka wola ze strony nas wszystkich, aby pomimo tego, co ustalimy teraz, co się wydarzy, na co osoby głuchonieme, niedosłyszące i słabo słyszące czekały, jednak te prace trwały szybciej i abyśmy szybciej doprowadzili do pełnej dostępności telewizji dla takich samych osób jak my. Dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł Urszula Pasławska, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na wstępie chciałam podziękować wnioskodawcom, ale również pani przewodniczącej podkomisji za przygotowanie i prowadzenie tego projektu ustawy, bo jest to ustawa oczywiście bardzo oczekiwana, bardzo potrzebna, bardzo ważna. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Europejskich Demokratów będzie popierał projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Proces, który ma zwiększyć dostęp osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu do programów telewizji publicznej oraz stacji komercyjnej, będzie przebiegać w sposób ewolucyjny. Tutaj właściwie ten projekt, który został złożony, i projekt, który wyszedł z komisji w jakimś sensie, znaczy, oczywiście nie jest tożsamy, dyskutowano na ten temat.

Dzisiaj jesteśmy - można to powiedzieć z niesmakiem - w ogonie Europy, jeśli chodzi o przepisy. Obecnie przepisy wymagają od nadawców dostosowania do potrzeb ludzi z niepełnosprawnościami jedynie 10% oferty. W polskiej telewizji w ten sposób nadawanych jest 18,5% programów, gdy średnia europejska to ok. 60%. Co więcej, to przede wszystkim seriale i powtórki programów rozrywkowych. Tymczasem ze środowisk osób z niepełnosprawnościami płyną sygnały, że znacznie bardziej zależy im na programach informacyjnych, wiadomościach i dziennikach. Jeszcze raz powtarzam, że nasz klub oczywiście popiera postulaty wskazane w ustawie. Są one zbieżne z zapisami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz polskiej konstytucji. Osoby z ograniczeniami, takimi jakimi są choroby narządu wzroku czy narządu słuchu, są przecież takimi samymi obywatelami i mają takie same nie tylko obowiązki, ale również prawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Zwiercan, Koło Poselskie Wolni i Solidarni. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania Komisji Kultury i Środków Przekazu o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Procedowana dziś nowelizacja ustawy ma na celu rozwiązanie problemu niedostępności programów telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzenie omawianej zmiany przyczyni się do zminimalizowania barier w dostępie do mediów, a także, co ważne, będzie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnościami. Nowelizacja przepisów ma na celu zobowiązanie nadawców programów telewizyjnych do zapewnienia dostępu do programów dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i dysfunkcją słuchu. Od 2024 r. co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programów ma posiadać udogodnienia umożliwiające odbiór osobom niepełnosprawnym. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że procedowany dziś projekt jest realizacją petycji, która trafiła do Senatu. Cieszę się, że zwykła obywatelska petycja nie została przeoczona i przerodziła się w inicjatywę ustawodawczą. Uważam, że omawiane dziś zmiany są zasadne i jak najbardziej potrzebne. Obecnie programy z udogodnieniami obejmują zaledwie 10% czasu antenowego. Proces zwiększenia liczby nadawanych programów z udogodnieniami musi zostać przeprowadzony jak najszybciej. Nie możemy zasłaniać się technicznymi czy finansowymi problemami z dostosowywaniem stacji telewizyjnych do emisji takich programów. Jak długo jeszcze osoby głuche, słabosłyszące czy niewidome mają czekać? Wszyscy bez wyjątku powinniśmy postawić się dziś na ich miejscu. My mamy pełny dostęp do wszystkiego, co nas otacza. Dlaczego więc osoby z niepełnosprawnościami nie otrzymują tego, co się im tak naprawdę należy? Dla nich to szansa na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, na rozwój. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. i systematycznie od tego roku rozszerzany ma być dostęp do udogodnień, aż do roku 2024, gdy co najmniej 50% czasu antenowego będzie posiadało udogodnienia dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i dysfunkcjami narządu słuchu. W petycji skierowanej do Senatu wnoszono, aby 100% kwartalnego czasu nadawanych programów posiadało takie udogodnienia. Uważam, że pełna dostępność programów z udogodnieniami powinna zostać zagwarantowana w krótszym czasie. Rozumiem jednak ograniczenia i dlatego mam nadzieję, że wejście w życie procedowanych rozwiązań będzie impulsem do dalszych zmian. Musimy robić, co tylko możliwe, by osobom z niepełnosprawnościami w Polsce żyło się dobrze, by nasz kraj był przyjazny dla nas wszystkich. Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za przyjęciem projektu ustawy. Dziękuję bardzo, pani poseł. Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Małgorzata Pępek. 1 minuta na zadanie pytania. Wysoka Izbo! Niezmiernie się cieszę, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wielu osób i że wejście zmienionej ustawy w życie, zgodnie z tym, co przegłosowano w trakcie prac komisji, będzie przyspieszone. Z drugiej strony szkoda, że ten projekt procedowany jest już od blisko roku. Zainteresowanych takimi zmianami jest obecnie około 4 mln osób wskazujących na wykluczenie społeczne, dyskryminację i łamanie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Do pana marszałka dotarła już chyba petycja w tej sprawie. W nowej wersji zmienianej ustawy mamy zobowiązanie do informowania o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji, które są dostępne dla niepełnosprawnych. I to też bardzo dobra i istotna zmiana. Chciałam zapytać, czy zostanie zagwarantowana osobom głuchym, słabosłyszącym i niewidomym [[Dzwonek]] dostępność programów o najwyższej oglądalności, napisy na żywo w „Wiadomościach” i programach publicystycznych. To dobra ustawa, która winna być zdecydowanie szybciej wdrażana. Czy nie można skrócić tego czasu? Bardzo proszę, pani poseł Halina Szydełko, klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Ten projekt mówiący o 50% to na pewno jest kompromis. Oczekiwania środowiska osób niepełnosprawnych są znacznie większe i na pewno słuszne. Moje pytanie dotyczy tych 50%, które teraz mamy zagwarantowane w projekcie ustawy. Czy w tych 50% będzie przewidziany procentowy udział poszczególnych programów informacyjnych, publicystycznych czy też materiałów filmowych, które będą objęte tymi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych? I czy przepisy wykonawcze, bo rozumiem, że tam powinno się to znaleźć, będą przewidywały taki podział? Bardzo proszę, pani poseł Joanna Fabisiak. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chodzi głównie o stwierdzenie, że to jest udogodnienie, gdy tymczasem można tu mówić o dostępności, o zwiększeniu dostępu do korzystania z dóbr kultury. Jeśli zajmujemy się tylko tą ustawą, to sytuacja wygląda nieźle, bo w ciągu roku będzie poprawa, w ciągu dwóch lat jeszcze większa.

Nie będę rozwijała tego wątku.

Zatem jeśli nawet nie możemy tego zapewnić w takim zakresie, jakbyśmy chcieli, przynajmniej nie używajmy języka dyskryminującego, języka obraźliwego często dla tych osób. One chcą, by mówić o tym, że to nie jest udogodnienie, tylko że to jest większy dostęp do korzystania z dóbr kultury. Bardzo proszę, pani poseł Zofia Czernow, Platforma Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Na pytania odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan minister Paweł Lewandowski.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

Oczywiście są kraje, w których jest to większe, ale można przyjąć, że 50% jest taką normą europejską i do takiej normy obecnie dążymy. Jako rząd zasadniczo popieramy projekt, który został przedłożony przez Senat, bo ten projekt uwzględnił także wszystkie poprawki zgłoszone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto zauważyć, że ministerstwo także przygotowywało taki projekt w ramach tzw. dużej ustawy czyszczącej, ustawy o radiofonii i telewizji, ale skoro ta inicjatywa została podjęta wcześniej przez Senat, to tylko poprosiliśmy o uwzględnienie uwag, które były zawarte w naszym projekcie rządowym. Czyli na pytania o procent w innych krajach i o możliwość, dlaczego 50%. 50% jest kompromisem, my ten kompromis na razie uważamy za wiążący, dlatego że nie nakłada zbytnich obciążeń na nadawców, a z drugiej strony jednak jest dużym krokiem naprzód. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle.

U nas zresztą nadawcy także do nas apelowali, żeby pozostawić to w kategorii samoregulacji, bo nadawcy oczywiście są odpowiedzialni i zdają sobie sprawę, ale wybraliśmy inną drogę. A więc poprawka, jak powtarzam, będzie rozpatrywana. Zobaczymy, jak się do niej odniesie cała komisja, jak się odniesie krajowa rada, która ma doświadczenie także chociażby z wprowadzaniem tego obecnego stanu prawnego. Gdyby się to udało, to ja -mogę tylko powiedzieć - osobiście byłabym w pełni szczęśliwa, aczkolwiek w tej chwili mamy 10%, a w przyszłym roku ma być 30%.

Prawda jest taka, jak powiedziałam, że ustawa to ramy. Wszystko będzie w rozporządzeniu, ale w dyspozycjach, jakie daliśmy krajowej radzie, jest wskazane, że w tym rozporządzeniu będzie mowa o rodzajach udogodnień w zależności od pory emisji, charakteru i rodzaju programu. Oczywiście to będzie musiało być w miarę szczegółowo rozpisane, ale nie zakończyła się rola odbiorców tych programów - oni w tej chwili muszą rozpocząć pertraktacje czy konsultacje z krajową radą i to trochę będzie zależało od tych rozmów. Ja o tym mówiłam, myśmy sobie doskonale zdawali sprawę z tego, że „udogodnienia” to jest takie słowo, które. Po prostu ktoś może oglądać program, i tyle. Niemniej były wysiłki ze strony krajowej rady, fachowców, ekspertów krajowej rady, którzy próbowali wyeliminować to słowo.

Pytanie: Co? Dziękuję oczywiście za uwagę i za uwagi.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń (druki nr 1996 i 2242) Bardzo proszę pana posła Andrzeja Matusiewicza o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń, druk sejmowy nr 1996. Marszałek Sejmu na 58. posiedzeniu Sejmu w dniu 6 lutego 2018 r. na podstawie art. 87 ust. 2 w związku z art. 90 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. Przypomnę, że projekt tej ustawy to projekt komisyjny, projekt Komisji do Spraw Petycji. Dotyczy on nowelizacji dwóch przepisów Kodeksu wykroczeń.

Dotychczasowy zapis był taki, że w tym art. 130 § 1 Kodeksu wyborczego był ujęty też art. 120, który dotyczy kradzieży drzewa z lasu czy przywłaszczenia tego drzewa, a art. 130 odnosił się do wyłączenia tych przypadków, jeśli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, materiały lub przyrządy wybuchowe, bo wtedy to nie jest wykroczenie, tylko jest to przestępstwo. A więc zasadne jest wyłączenie z tego przepisu art. 120 Kodeksu wykroczeń, który - jak już powiedziałem - dotyczy kradzieży drzewa. Jego dotychczasowe brzmienie było takie: „Kto prowadzi zakład opieki zdrowotnej lub zakład leczniczy dla zwierząt bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny” Termin „zakład opieki zdrowotnej” został wyeliminowany z obrotu prawnego ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, gdyż wprowadzono nowe pojęcie podmiotu leczniczego.

Utrzymano art. 2 tego projektu, czyli minimalny termin wejścia w życie ustawy 14 dni od ogłoszenia. Wnoszę o przyjęcie tego projektu w imieniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w sposób niezmienny popiera przedmiotowy projekt. Nowelizacja Kodeksu wykroczeń jest tutaj konieczna. Jest to zmiana, nowelizacja czyszcząca, czyli tak naprawdę eliminująca sprzeczności, które z przepisów wynikają. W pierwszym wypadku jest to ewidentna nieprawidłowość, natomiast w drugim wypadku jest to nieaktualny przepis w związku ze zmianą innych merytorycznych przepisów. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera proponowane zmiany, po wniesionych też korektach ze strony komisji. Bardzo proszę, pani poseł Katarzyna Osos, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo! Klub Platforma Obywatelska tak jak podczas pierwszego czytania, tak również po pracach w komisji popiera projekt. Jak już tu zostało wcześniej powiedziane, nie budzi on kontrowersji, jest czyszczący, eliminuje przepisy, które nie spełniają zasad prawidłowej legislacji, również wprowadzone podczas prac komisji poprawki są zasadne i Platforma Obywatelska będzie popierać projekt. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł.

Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, druk nr 2286 i 2314. Projektowana ustawa zawiera zmiany nie tylko umożliwiające zgodność przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej, ale także wprowadza inne modyfikacje niezwiązane z koniecznością dostosowania do przepisów unijnych. Dodatkowo należy wskazać, że niektóre z proponowanych regulacji zawartych w projektowanej ustawie mają na celu wypełnienie zobowiązań nałożonych przez Komisję Europejską m.in. w związku z trwającym procesem notyfikacji publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne w 2015 r. na restrukturyzację. Projektowana ustawa wprowadza uzupełnienie w art. 22 w zakresie zasad bezpośredniego zawierania umów, dodaje nowy art. 22b przyznający organizatorowi prawo do podjęcia negocjacji z podmiotem, który jako jedyny wyraził zainteresowanie udziałem w procedurze przetargowej bez konieczności ponownej publikacji ogłoszenia przetargu, oraz wprowadza uzupełnienie w art. 49 ustawy poprzez poszerzenie zakresu informacji przekazywanych przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego marszałkowi województwa, który zobowiązany jest do przygotowania informacji zbiorczej dotyczącej publicznego transportu zbiorowego z podziałem na transport autobusowy i kolejowy, oraz nałożenie obowiązków sprawozdawczych dodatkowo na związki powiatowo-gminne, związki metropolitalne i marszałków województw. Ponadto projektowana ustawa zawiera m.in. umożliwienie zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych w przypadku powierzenia ich wykonywania temu samemu operatorowi. Na skutek uwag zgłoszonych podczas konsultacji międzyresortowych projektodawca zdecydował się, że zapisy dotyczące przewozów pasażerskich pomiędzy stacjami ulokowanymi w sąsiednich województwach zostały usunięte z obecnie projektowanej ustawy. Rozwiązanie tej bardzo ważnej kwestii nastąpi w innym projekcie, w którym zostaną wypracowane przejrzyste rozwiązania problemu połączeń stykowych. Podsumowując, w projektowanej ustawie o publicznym transporcie zbiorowym proponowane rozwiązania nie wywołują skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Projekt ustawy jest zgodny z prawem unijnym, a rozwiązania zawarte w projekcie nie będą miały wpływu na działalność mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Klub Prawa i Sprawiedliwości w pełni popiera projektowaną ustawę o publicznym transporcie zbiorowym i będzie głosował za jej przyjęciem. Bardzo proszę, pan poseł Stanisław Lamczyk, Platforma Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma na celu zapewnienie zgodności przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Dokładnie chodzi o rozporządzenie Unii Europejskiej z roku 2016 nr 2338, które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, a które weszło w życie dnia 24 grudnia 2017 r. W uzasadnieniu postuluje się, żeby projektowana ustawa weszła w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Jest to oczywiście niezrozumiały pośpiech, ponieważ 20 października 2016 r. na tej sali mówiliśmy o projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym i wtedy sygnalizowane były pewne problemy, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w kontekście uchwalenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

Są to, można powiedzieć, wytyczne dla ministra, który w drodze rozporządzenia określi minimalny zakres informacji publikowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dokumentach koncesji dotyczących minimalnego okresu pomiędzy ogłoszeniem o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego a rozpoczęciem świadczenia usługi oraz minimalnego okresu pomiędzy zawarciem umowy o świadczenie usługi a rozpoczęciem świadczenia usługi, warunków dostępu do taboru kolejowego niezbędnego do realizacji usługi, danych dotyczących rynku, na którym ma być świadczona usługa, w tym przychodów oraz wymagań wobec systemów taryfowo-biletowych, obowiązki w zakresie gwarancji socjalnych i zasad przyjmowania pracowników, mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystości procedury wyboru operatora oraz zabezpieczenia odpowiednich warunków realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Pozwolę sobie na ręce pani marszałek przekazać treść tej poprawki. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana posła Mirosława Suchonia, klub

Projekt zapewnia przede wszystkim możliwość kontynuacji tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli działalności prowadzonej na podstawie wpisu do CEIDG, po śmierci przedsiębiorcy.

I co jest też ciekawe, a jednocześnie ważne z punktu widzenia potrzeby wprowadzenia omawianej regulacji, tę formę działalności wybiera ciągle ok. 80% początkujących firm także dzisiaj.

Firma prowadzona jednoosobowo jest dzisiaj - i to jest ten problem, na który odpowiadamy - nierozerwalnie związana z jej właścicielem. Śmierć przedsiębiorcy powoduje, że kończy się także byt prawny przedsiębiorstwa, a wiemy, że czasami są to firmy budowane latami, często nakładem pracy już nie tylko samego przedsiębiorcy, ale także jego rodziny, jego współpracowników, czyli, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, firma dzisiaj umiera wraz z jej właścicielem.

W praktyce śmierć przedsiębiorcy oznacza, że nie można wykonywać, kontynuować wielu kontraktów handlowych, jej skutkiem jest także wygaśnięcie umów o pracę, nie można posługiwać się NIP-em zmarłego przedsiębiorcy, co jest też oczywiście równoznaczne z tym, że nie ma płynności rozliczeń podatkowych, wygasają decyzje administracyjne typu koncesje, licencje, zezwolenia, co też często jest wręcz niezbędne do funkcjonowania firmy, wreszcie brak jest dostępu do rachunku bankowego prowadzonego na potrzeby przedsiębiorstwa. Praktyka obrotu pokazuje, że do zakończenia formalności spadkowych, które często trwały wiele miesięcy, a czasami nawet w lata to przechodziło, następcy prawni mają trudności z bieżącym zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Dla takiej firmy już nie ma tak naprawdę powrotu na rynek.

Bo osoby, które zakładały swoje firmy w okresie transformacji gospodarczej, ustrojowej, dzisiaj zbliżają się do wieku dojrzałego lub ten wiek już osiągnęły. Sprawdziliśmy w CEIDG, że dzisiaj mamy 212 tys. przedsiębiorców, którzy ukończyli 65. rok życia, i w ciągu ostatniego roku ta liczba wzrosła aż o 15 tys.

Myślę, że ważne i godne podkreślenia jest to, że prace nad tym projektem rozpoczęły się z inicjatywy firm rodzinnych, i to ich sygnalizacja sprawiła, że ministerstwo podjęło się uregulowania tego zagadnienia. Ważne dla nas w trakcie procesu legislacyjnego było to, że aktywność firm pozwoliła nam podchodzić do pewnych praktycznych problemów właśnie w konsultacji z nimi, kiedy zastanawialiśmy się nad jakimiś praktycznymi, licznymi dylematami, bo to jest trudna ustawa.

Ale z punktu widzenia globalnego firmy rodzinne stanowią dzisiaj ok. 35% polskich przedsiębiorców, wytwarzając ok. 10% PKB, i w sektorze przedsiębiorstw zatrudniają ok. połowy pracowników.

Tak więc proponowane przez nas rozwiązania umożliwiają płynną kontynuację działalności firmy po śmierci przedsiębiorcy, osoby fizycznej.

Taką instytucją, która służy utrzymaniu czy realizacji celu, jest przede wszystkim instytucja zarządu sukcesyjnego.

Zarządca będzie także występował w postępowaniach cywilnych, administracyjnych, podatkowych związanych z przedsiębiorcą, będzie mógł dochodzić wierzytelności zmarłego przedsiębiorcy, będzie mógł spłacać należności, tak że spadkodawca będzie mógł uzyskać interpretacje podatkowe. Będzie to wszystko to, co wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem, w tym również dostęp do firmowych rachunków bankowych, co dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, w zasadzie jest przecięte w momencie śmierci przedsiębiorcy. Korzystanie z rozwiązań oczywiście będzie w pełni dobrowolne. To od samego przedsiębiorcy, a po jego śmierci od jego sukcesorów będzie zależało, czy dojdzie do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego i instytucji zarządu sukcesyjnego.

Do powołania zarządcy sukcesyjnego wystarczy pisemne oświadczenie przedsiębiorcy, zgoda zarządcy na pełnienie tej funkcji i wpis zarządcy do CEIDG.

Rozwiązanie polegające na możliwości ustanowienia prokury przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG przewidzieliśmy ostatnio w pakiecie tzw. konstytucji biznesu.

Też różnego rodzaju badania pokazują, że wielu przedsiębiorców o tym nie myśli, a przynajmniej nie przewiduje tych kroków po swojej śmierci.

Bo tutaj łączymy przepisy cywilne, typu: spadkowe, zobowiązaniowe, proceduralne, czyli z k.p.c., prawo administracyjne, prawo publiczne, prawo podatkowe.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Szanowna Pani Marszałek! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z druku nr 2293. Ogólnie rzecz ujmując, projekt dotyczy wprowadzenia zmian legislacyjnych, które ułatwiałyby dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa osoby fizycznej wpisanej do CEIDG na analogicznych zasadach jak za życia przedsiębiorcy w okresie, co do zasady, między otwarciem spadku a jego działem. Działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne to zdecydowanie najbardziej popularna forma wykonywana przez ponad 3 mln osób zarejestrowanych w systemie REGON oraz ponad 300 tys. spółek cywilnych. Najważniejszymi cechami charakteryzującymi firmy rodzinne są: budowanie przedsiębiorstwa na własności, sukcesja rodzinna oraz zaangażowanie rodziny w prowadzenie biznesu. Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed firmami rodzinnymi jest kwestia sukcesji pokoleniowej. W obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy de facto kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Wiąże się z tym szereg problemów dotyczących sfery prawa prywatnego, jak również publicznego, które w praktyce utrudniają kontynuację czy wznowienie działalności przedsiębiorczej przez następców prawnych. Do najważniejszych z nich należą: brak ośrodka decyzyjnego, jednej osoby uprawnionej do prowadzenia spraw przedsiębiorcy i samodzielnej reprezentacji wszystkich następców prawnych, ograniczone możliwości posługiwania się choćby tymczasowo firmą przedsiębiorcy, wygaśnięcie umów zawartych przez przedsiębiorcę, wygaśnięcie decyzji administracyjnych niezbędnych do prowadzonego rodzaju działalności gospodarczej, takich jak koncesje, licencje czy pozwolenia, oraz chociażby trudności z dostępem do rachunku bankowego. Tak że w aktualnym stanie prawnym zachowanie pełnej ciągłości działalności gospodarczej jest w praktyce niemożliwe. Podobna sytuacja dotyczy prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w formie spółek cywilnych. Śmierć wspólnika niejednokrotnie powodować może zagrożenie dla istnienia spółki, szczególnie tej dwuosobowej. Podstawowym celem regulacji jest zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków do zachowania ciągłości przedsiębiorstwa po ich śmierci. Dodatkowym celem regulacji jest wzmocnienie praw osób trzecich związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim pracowników, kontrahentów, konsumentów i innych podmiotów współpracujących z przedsiębiorstwem. Dzięki kontynuacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, które będzie w dalszym ciągu generować zyski, zachowane zostaną miejsca pracy, zwiększą się szanse na dalszy rozwój przedsiębiorstwa budowanego niekiedy osobistymi staraniami przedsiębiorcy i członków jego rodziny czasami przez wiele lat. Wprowadzenie do porządku prawnego rozwiązań umożliwiających kontynuację funkcjonowania przedsiębiorstwa osoby fizycznej po jej śmierci będzie wymagało wprowadzenia do systemu prawa nowej ustawy kompleksowo regulującej funkcjonowanie przedsiębiorstwa w okresie tzw. zarządu sukcesyjnego, jak również obejmie zmianę szeregu ustaw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy czy prawa podatkowego. Ustawa ta jest bardzo oczekiwana przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także - i przede wszystkim - przez ich rodziny. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera projekt tej ustawy i jest za skierowaniem go do dalszych prac w komisji. Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Cel tego projektu, który jest tutaj dzisiaj przedstawiany, jest bardzo ważny, ponieważ projekt ma zapewnić, by przedsiębiorstwo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie kończyło bytu prawnego wraz ze śmiercią tej osoby. Ten cel jest bardzo ważny z uwagi na jeszcze inne aspekty, które dodam, a mianowicie powinien to być system powszechny, powszechnie stosowany, tak by nie tracili na tym właściciele, by nie tracili na tym pracownicy i by nie tracił na tym oczywiście obrót gospodarczy. Te dwie instytucje, o których tutaj pan minister wspomniał, instytucja zarządu i zarządcy sukcesyjnego, mają to zagwarantować.

Obecnie środowiska przedsiębiorców właśnie oczekują lepszego rozwiązania, ponieważ obecne testamentowe przekazywanie, z którego można było korzystać, jednak w bardzo minimalnym stopniu jest wykorzystywane przez przedsiębiorców, a to znaczy, że oprócz tej funkcji, o której powiedziałam, ta funkcja edukacyjno-informacyjna jest bardzo istotna. Dlatego tak ważna jest świadomość prawna osób fizycznych, przedsiębiorców oraz ich rodzin i oby ta ustawa spowodowała i wymusiła tę świadomość. W pracach w komisji oczywiście będziemy poprzez propozycje, pytania czy głębsze debaty nad tym starali się wesprzeć tę ustawę, tak aby ona ten swój cel mogła spełnić. Istotne jest tutaj rozwiązanie również tego powołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy. Pan minister to dość dokładnie wyjaśnił.

W tym krótkim czasie osoby, które są uprawnione do tego, by powołać zarządcę, czyli małżonek przedsiębiorcy, osoba, która przejęła zapis windykacyjny czy spadkobierca, będą musiały uzyskać zgodę wszystkich osób, które mogą mieć wpływ na tego zarządcę.

Problemem jest też w mojej ocenie to, że w tak krótkim czasie trzeba podjąć decyzję o przyjęciu spadku czy o przyjęciu zapisu windykacyjnego. Tak że te ramy czasowe na pewno powinniśmy bardzo szczegółowo przeanalizować i zastanowić się nad tym, czy one nie powinny być tutaj inaczej uregulowane. Bardzo ważne jest też to, żeby te osoby, które są uprawnione do powoływania zarządcy, miały świadomość, jakie on będzie wykonywał zadania, jaką będzie ponosił w związku z tym odpowiedzialność i jakie też skutki tego będą ciążyły na tych osobach powołujących zarządcę.

Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na art. 21 i 22, a także na relacje między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą i na to, o czym powiedziałam, na odpowiedzialność za zobowiązania i wszystkie podejmowane w tym czasie decyzje. Chodzi tu również o kwestię decyzji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, które nie wygasną, jeśli w terminie 3 miesięcy ten zarządca złoży stosowny wniosek i oświadczy, że przyjmuje warunki wskazane w decyzji i będzie jeszcze oczywiście te warunki spełniał. Tutaj również ten czas 3 miesięcy wydaje się zbyt krótki, więc w tej kwestii będziemy próbowali przedstawić swoje propozycje. Jesteśmy za tym, aby przekazać ten projekt do dalszych prac w komisji.

Dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Cieszy mnie to, że wnioskodawca zajął się tym trudnym, ale bardzo ważnym z punktu widzenia przedsiębiorców problemem. Jak dobrze wiemy, jeśli przedsiębiorstwo nie funkcjonuje, nie ma wpływów podatkowych, ale jest to też rzeczywisty problem. Zacznę więc od pozytywów tej ustawy. Przede wszystkim ustawa zapewni ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstw po śmierci przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobową, wzmocni ochronę osób trzecich związanych z przedsiębiorstwem, szczególnie pracowników, których umowy o pracę obecnie wygasają w chwili śmierci i w zasadzie Kodeks pracy nie chroni ich tak samo jak osób zatrudnionych w spółkach czy w innych formach działalności gospodarczej. Natomiast są też w tej ustawie mankamenty i kontrowersje, które, mam nadzieję, uda się rozwiązać podczas prac w komisji. Rzeczywiście może być to trudne w sytuacji dłuższych postępowań spadkowych. Innym problemem jest ograniczenie skutków podatkowych wyłącznie do firm jednoosobowych. Brak jest bardziej kompleksowego podejścia do zagadnienia i objęcia regulacją wszystkich sytuacji, w których do chwili śmierci dana osoba uzyskiwała dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Moim zdaniem jednak największym problemem, który, mam nadzieję, uda się rozwiązać, jest brak przepisów umożliwiających jednoosobowemu przedsiębiorcy przekształcenie działalności w spółkę osobową, np. w spółkę jawną z udziałem członków jego rodziny. Wprowadzenie takich przepisów umożliwiających jednoosobowym przedsiębiorcom przekształcenie działalności także w spółkę osobową spowodowałoby, że w przypadku śmierci jednego ze wspólników przedsiębiorstwo miałoby możliwość bezproblemowego kontynuowania swojej działalności na takich samych zasadach jak dotychczas. Tak że ustawa jest dobra. Mam nadzieję, że w trakcie prac w komisji uwzględnione zostaną uwagi przedstawione tutaj, na sali plenarnej, przede wszystkim te dotyczące stworzenia możliwości przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę osobową prawa handlowego, co od dawna postulują przedstawiciele przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jerzy Meysztowicz, klub Nowoczesna. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Jak już tu wcześniej powiedziano, sprawa sukcesji firm jednoosobowych jest poważnym, realnym problemem przedsiębiorców. W obecnym stanie prawnym sukcesja firmy rodzinnej jest możliwa, ale skomplikowana i wymaga wcześniejszych przygotowań, których większość przedsiębiorców niestety nie czyni. Ponadto przekazanie firmy w testamencie w formie tzw. zapisu windykacyjnego wymaga zapłacenia podatku od spadku, co może poważnie ograniczyć możliwości i chęci przyjęcia biznesu przez sukcesora. Stąd w momencie śmierci przedsiębiorcy pojawiają się problemy z dalszym prowadzeniem firmy, często prowadzące nawet do upadłości. Wygasają wszystkie umowy, w tym umowy o pracę. Spadkobiercy nie mogą nawet tymczasowo posługiwać się m.in. nazwą firmy czy NIP-em zmarłego przedsiębiorcy, a nawet nabywając w spadku składniki majątkowe tego przedsiębiorstwa, nie nabywają praw niematerialnych z tym związanych. Tracą na tym i spadkobiercy, i gospodarka jako całość. Problematyczne jest też zarządzanie przedsiębiorstwem w trakcie wielomiesięcznych postępowań spadkowych.

W okresie do powołania zarządu sukcesyjnego małżonek spadkobierca może wykonywać czynności niezbędne do zachowania majątku i możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa, w szczególności zaspokajania wymaganych roszczeń, przyjmowania należności i sprzedaży aktywów obrotowych.

Generalnie ujmując, uważamy, że rzeczywiście ta ustawa jest potrzebna. Ona powinna zostać uchwalona już wcześniej, dlatego że wiele małych firm niestety upadło - nie można było kontynuować działalności, dlatego że rzeczywiście po śmierci właściciela tak na dobrą sprawę firma przestawała istnieć. Mianowicie zwolnienie z podatku od spadku obowiązuje w przypadku kontynuacji działalności przez 5 lat, nawet gdy dalsze działanie przedsiębiorstwa nie ma uzasadnienia ekonomicznego lub ogłoszona zostanie upadłość.

Rekomendacja Nowoczesnej jest taka, aby dalsze prace nad tą ustawą odbywały się w komisji. Bardzo proszę, pan poseł Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów mam zaszczyt zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie. Czuję, że pan minister tutaj bardzo szczegółowo przedstawił uzasadnienie potrzeby uchwalenia takiej ustawy.

Wszyscy wiemy, jak trudne są podziały majątku, sprawy związane z masą upadłościową, załatwieniem roszczeń poszczególnych członków rodziny. To powoduje, że przedsiębiorstwo w tym czasie może całkowicie upaść, zostać zlikwidowane. Stracą nie tylko właściciele, nie tylko spadkobiercy, ale również pracownicy, którzy są tam zatrudnieni. Dobrze, że rząd podjął się takich prac.

Nie będę tutaj mówił o uwagach do tej ustawy, bo myślę, że te uwagi będziemy zgłaszać na posiedzeniu komisji czy podkomisji. Myślę, że jeszcze wiele zmian tam się znajdzie, bo tak jak pan minister powiedział, przez 2 lata pracował pan nad tą ustawą, więc widać, że sprawy są poważne i wymagają wielu uzgodnień, i tak prawdopodobnie będzie w komisji. W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Europejskich Demokratów wnioskuję o dalsze prace w komisjach. Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zadać pytanie? Jeżeli nie, zamykam listę. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Paweł Bańkowski, Platforma Obywatelska. Czas na zadanie pytania - 1 minuta. Panie Ministrze!

Tymczasem wpis do CEIDG nie przesądza o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej, stanowi jedynie podstawę rozpoczęcia działalności gospodarczej w rozumieniu jej legalizacji i nie jest zdarzeniem utożsamianym z podjęciem takiej działalności. Pytanie, panie ministrze: Dlaczego zakres podmiotowy projektowanej ustawy nie obejmuje osób fizycznych, które w momencie swej śmierci faktycznie wykonywały we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a więc będących w chwili śmierci przedsiębiorcami w rozumieniu Kodeksu cywilnego mimo braku ich wpisu CEIDG? Czy takie brzmienie projektowanej ustawy jest zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej? Zgodnie z brzmieniem ustawy od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Czy celem autorów projektowanej ustawy [[Dzwonek]] jest utrzymanie w mocy umów zawartych przez zmarłego przedsiębiorcę przed jego śmiercią? Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Pępek, Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo! Ministerstwo rozwoju chce, by mimo śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą była zachowana ciągłość rozliczeń podatkowych związanych z tą działalnością. Projekt w ocenie wielu przedsiębiorców jest niedopracowany. Pojawiły się nawet złośliwe komentarze i pomysły, żeby przedsiębiorca, zanim uda się na drugi świat, swoją zadłużoną działalność zapisał w spadku państwu polskiemu. Dziedziczenie nie obejmuje praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych, w przypadku wielu zezwoleń nie ma możliwości przejęcia decyzji przez następcę, więc ciągłość funkcjonowania biznesu będzie zahamowana dla spadkobierców z chwilą śmierci przedsiębiorcy. W konsekwencji dochodzi do tego, że następca nie będzie mógł prowadzić działalności lub wykonywać określonych czynności, dopóki nie uzyska stosownych decyzji na swoją rzecz.

Dziękuję bardzo. Proszę, pan poseł Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska. Nie ma pana posła. Pan poseł Zbigniew Gryglas, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Jest ona korzystna nie tylko dla przedsiębiorstw rodzinnych, które będą mogły kontynuować działalność, ale także dla całej gospodarki. Trudno przecenić to znaczenie.

Pytanie: Dlaczego tego typu regulacja nie znalazła się w projekcie? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Maria Małgorzata Janyska, Platforma Obywatelska. Czy jest potrzeba potwierdzania możliwości wykonywania decyzji związanych z przedsiębiorstwem? Jeśli to nie są decyzje, które dotyczą, bo te są wyłączone, indywidualnie, osobowo właściciela, a są to licencje, są to koncesje czy zezwolenia, to gdyby np. przedsiębiorca żył i powierzył zarządzanie swoją firmą menedżerowi czy dyrektorowi, obojętnie, jak to nazwie, jak to jest w strukturze organizacyjnej, nie musiałby tego potwierdzać, więc pytanie, czy tutaj ten aspekt jest niezbędny. Drugie pytanie.

Panie Ministrze!

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Panie ministrze, jaka jest sugestia ministerstwa, do której komisji trafi ta ustawa? Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze! Mam też krótkie pytanie o terminy.

Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź na pytania przedstawiciela wnioskodawców podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii pana ministra Mariusza Haładyja. Bardzo proszę. Pani Marszałek!

Po pierwsze, nie ma informacji, że one w ogóle prowadziły działalność gospodarczą. Czy w związku z tym powinniśmy prowadzić, czy organy państwa powinny prowadzić jakieś postępowania wyjaśniające, gdy ta działalność była prowadzona, ale niezarejestrowana?

Drugie pytanie dotyczyło tego, czy utrzymujemy kontrakty cywilne, jak rozumiem, czyli handlowe.

Pani poseł Pępek stwierdziła, że nie dopracowaliśmy projektu, bo są decyzje administracyjne, które wygasają, w związku z tym jest jakaś ogromna dziura, jak rozumiem, w tym projekcie, gdyż on tego nie przewiduje.

Oczywiście działania informacyjne będą musiały się odbyć i oczywiście powoli o nich myślimy, tylko wcześniej chcielibyśmy też wiedzieć, że ustawa uzyska akceptację najpierw parlamentu, a później prezydenta. Jeżeli tak się stanie, to mamy przewidziany pewien pakiet działań.

Pan poseł Gryglas pytał, dlaczego nie ma przekształcenia w spółkę, zresztą też jeden z posłów o to pytał w trakcie prezentowania stanowisk klubów.

W ogóle polski system prawa nie zna czegoś takiego jak jednoosobowa spółka osobowa. Jest jedynie ten roczny okres prowadzenia w takiej formule spółki partnerskiej po śmierci jednego z dwóch partnerów takiej spółki, natomiast generalnie nie przez przypadek polski system prawa takiej instytucji nie przewidział. Tak naprawdę przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę osobową w zasadzie byłoby moim zdaniem chyba powołaniem nowego bytu prawnego, czyli spółki osobowej.

Wycofanie się z ograniczeń - mam wrażenie, że to jest pytanie wykraczające poza dzisiejszą dyskusję. Zwykły. Aha, pan poseł Kasprzak pytał, jakich czynności nie będzie mógł wykonywać zarządca sukcesyjny.

To jest oczywiście pewnego rodzaju dylemat i nie ukrywam, że mamy jakiś wzór matematyczny, który nam pozwolił wyliczyć, że 2 miesiące to jest optimum.

Szybciutko kończę.

Bo co się dzieje w ciągu tych 2 miesięcy? Kontrahent też żyje w jakimś sensie w stanie niepewności. W stanie niepewności żyją także pracownicy, czy będzie powrót tej firmy, czy go nie będzie, czy mają szukać nowej roboty, czy liczyć, że spadkobiercy podejmą tę kwestię. Mamy też stan zawieszenia, jeśli chodzi o decyzje administracyjne, mamy kwestię przywrócenia NIP-u.

Z naszej perspektywy to wydaje się... tzn. to nie jest jakiś gigantyczny problem.

Mam przyjemność zaprezentować projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Jesteśmy w 24. roku funkcjonowania tego mechanizmu.

A zatem projektowane regulacje stanowią z jednej strony odpowiedź na zmiany społeczne i gospodarcze, jakie zachodzą nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, oraz są odpowiedzią również na założenia wpisane w „Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, średniookresową strategię, w której również pewne zasady i założenia dotyczące przyciągania nowych inwestycji czy też wspierania nowych inwestycji zostały zdiagnozowane. Jednym z zakładanych efektów „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” jest trwały rozwój gospodarczy, to po pierwsze, a po drugie, rozwój zrównoważony terytorialnie.

Po pierwsze, analizy nie są jednoznaczne.

I tak widzimy, pomimo iż przy wschodniej ścianie Polski mamy specjalne strefy ekonomiczne, że ilość zainteresowanych podmiotów inwestowaniem tam nie dorównuje w żaden sposób ilości tych, którzy są zainteresowani inwestowaniem przy granicy zachodniej czy też na terenach, które dzisiaj i tak są w dobrym stanie rozwojowym, jeżeli chodzi o wskaźniki makroekonomiczne.

Wprowadzenie mechanizmów, które istotnie poprawią jakość i ilość inwestycji na tych białych plamach na mapie Polski rozwojowej, szczególnie nas tutaj interesowało. Dlatego zaprojektowany w ustawie system wsparcia w postaci prawa do uzyskania przez przedsiębiorcę zwolnienia od podatku dochodowego stanowić będzie ważne i skuteczne narzędzie zachęcające przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju. Tak jak państwo posłowie zapewne pamiętają, projekt ten przedstawialiśmy tak: cała Polska specjalną strefą ekonomiczną. Co się zatem zmienia w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów? Po pierwsze, w kryteriach oceny inwestycji, które będą mogły liczyć na uzyskanie przywileju strefowego, stawiamy na rozwój innowacyjnych dziedzin działalności gospodarczej.

Zatem raczej jakość tej inwestycji jest tym, co chcielibyśmy w procesie przyznawania przywileju oceniać. Kolejny nie mniej istotny element to tworzenie nowych stabilnych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jeśli mówmy, że jednym z celów SOR-u jest zrównanie dochodów pracowników wykwalifikowanych, polskich pracowników z pracownikami w starych państwach członkowskich Unii Europejskiej, to z całą pewnością lokowanie wysokowolumenowych, wysokowartościowych przemysłów przetwarzających znajdujących się wysoko w łańcuchu wartości jest tym, co chcemy nagradzać przywilejem strefowym. Zależy nam na tworzeniu dzięki temu mechanizmowi nowych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz na ich wykorzystaniu w gospodarce, zwiększeniu konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług, rozwoju eksportu, dalszym rozwoju eksportu, bo przypomnę, że te wskaźniki za I kwartał również są dla nas bardzo optymistyczne.

Te specjalne strefy ekonomiczne, które zostały utworzone 20 lat temu, takim zmianom nie były przez te 20 lat poddawane.

W przeciwieństwie do dotychczasowego systemu przedsiębiorca będzie mógł starać się o ulgę na dowolnym terenie, na którym można prowadzić działalność gospodarczą. Spółka strefowa dzisiaj nie będzie się w pierwszej kolejności zajmować poszerzaniem swoich terenów, a następnie ich zbywaniem, jak to dotychczas miało miejsce, ale ma się zająć przede wszystkim profesjonalną obsługą inwestora, który wybiera sobie.

Natomiast rzeczywiście inwestor będzie miał większą swobodę w wyborze. Co to również implikuje w praktyce? Dzisiaj jest tak, że specjalna strefa ekonomiczna występuje o zgodę na nabycie terenu, następnie ta zgoda często jest okupiona oczywiście dyskusją, w zależności od planu zagospodarowania przestrzennego, z organami samorządu lokalnego, z agencją nieruchomości.

Ustawa wyeliminuje także sytuację, w której niektóre powiaty nie były objęte obszarem strefy ekonomicznej, a inne miały kilka stref działających na ich terytorium. Ustawa ta, aby było jasne, nie zwiększa biurokracji, ponieważ nie ulegnie zwiększeniu liczba spółek obsługujących inwestorów, spółki dostaną nowe zadania - te spółki, które funkcjonują już dzisiaj. Będą, po pierwsze udostępniać przedsiębiorcom na podstawie umowy składniki mienia, których zarządzający jest właścicielem. Będą prowadzić działania promocyjne na rzecz podmiotów działających na terenie strefy. To też jest pewna zmiana wektora. Spółki zajmowały się przede wszystkim przyciąganiem i osadzeniem inwestycji na swoim terenie. Dzisiaj będziemy w myśl ustawy wymagać od stref również ich aktywnego wsparcia proeksportowego, wychodzenia na zewnątrz z produktami i usługami wypracowywanymi przez firmę. Cały pakiet informacyjny dotyczący informacji o rynku pracy, pośredniczenie pomiędzy inwestorem a powiatowymi urzędami pracy, jeśli chodzi o zasób kadr niezbędnych dla danego sektora, dla danego przedsiębiorcy. Wreszcie współpraca w kształceniu, w tworzeniu rozwiązań do kształcenia na potrzeby firm działających w obszarze, w jurysdykcji specjalnej strefy ekonomicznej.

Chcielibyśmy, aby taka mapa pojawiła się jak najszybciej, bo istotnie taką mapą dzisiaj nigdzie żaden organ ani żadna instytucja w Polsce nie dysponują. Zarządzający obszarami strefowymi będą wykonywali swoje zadania na podstawie sporządzonego przez siebie planu rozwoju inwestycji.

Co będzie warunkowało decyzję o wsparciu? Podstawą udzielania pomocy będzie otrzymanie przez potencjalnego inwestora decyzji o wsparciu. Decyzja ta będzie określać okres jej obowiązywania, tak jak to ma miejsce i dziś w specjalnych strefach ekonomicznych, a co za tym idzie, okres, przez jaki przedsiębiorca będzie uprawniony do skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku dochodowego.

Ta decyzja będzie wydawana na okres od 10 do 15 lat, a na terenach, które do wejścia w życie ustawy były włączone w strefy ekonomiczne, decyzja będzie wydawana na okres 15 lat.

Ustawa przewiduje dwojaką ocenę inwestycji. Po pierwsze, będziemy oceniać je przez pryzmat wysokości nakładów inwestycyjnych - to, o czym mówiłam wcześniej, że wolumen inwestycji jest istotny. Próg nakładów będzie inny w zależności od wielkości firmy i poziomu rozwoju powiatu. Co to oznacza?

To też, przypomnę, jeden z naszych celów, nie tylko ilość małych i średnich firm, z których jesteśmy bardzo dumni w Polsce, jeśli chodzi o wkład małych i średnich firm do PKB, ale także ilość zatrudnianych pracowników. Natomiast jednym z celów, również bardzo istotnych, jest to, aby te małe firmy stawały się średnimi, a średnie - dużymi. Wierzymy w to, że udostępnienie małym i średnim firmom możliwości skorzystania z dodatkowych przywilejów, jakie daje mechanizm strefowy, pozwoli im szybciej urosnąć. Zgodnie z art. 28 również tworzy się ewidencję wsparcia inwestycji, której celem będzie pozyskanie danych wykorzystywanych do obsługi procesu inwestycyjnego, przeprowadzenia analiz w zakresie efektów funkcjonowania wsparcia udzielanego na podstawie niniejszej ustawy.

To ona będzie takim stałym monitoringiem tego i da też łatwość dostępu do oceny tego, w jaki sposób realnie ten mechanizm strefowy działa i wpływa na polską gospodarkę. Ewidencja będzie obsługiwana przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

One mają zapewnione i zagwarantowane warunki, na których dzisiaj pracują, bo ta ustawa takie przyjmuje założenia. Dla tych przedsiębiorców, bo przecież proces nie jest zatrzymany w biegu.

A zatem stabilność warunków prowadzenia działalności to jedna rzecz. Kolejna rzecz to stabilne zatrudnienie.

Trzecia istotna rzecz to jest kwestia odpowiedzialnego rozwoju, o którym mówimy, odpowiedzialnego, czyli zrównoważonego terytorialnie. I piąta to nadzieja na szybki rozwój technologii innowacyjnych, nowoczesnych, tych, które są napędem globalnej gospodarki. Mam nadzieję, że ten projekt spotka się z państwa zainteresowaniem. Dziękuję, pani minister. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Ewa Malik z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić opinię odnośnie do projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, druk poselski nr 2307. W polskim ustawodawstwie istnieje ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, zwana ustawą o SSE, uchwalona 20 października 1994 r., która reguluje kwestie wynikłe z konieczności pobudzania inwestycji, jednocześnie z procesem likwidacji wysokiego bezrobocia strukturalnego, którego tak wysoki poziom w latach 90. był skutkiem przemian ustrojowych po 1989 r. Obecnie duża liczba przedsiębiorstw stara się uzyskać zwolnienie od podatku dochodowego, a zainteresowanie tą formą pomocy od państwa wzrasta. Na koniec 2016 r. liczba ważnych zezwoleń na prowadzenie na terenach SSE działalności gospodarczej to 2263, skumulowana wartość zainwestowanego kapitału wyniosła ok. 112 mld zł, a liczba zatrudnionych dzięki tym inwestycjom pracowników wyniosła ponad 332 tys. Te fakty przemawiają niezbicie za koniecznością utrzymania narzędzi państwa opartych na ulgach podatkowych dla przedsiębiorców deklarujących realizację nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy, przy czym instrument zwolnień podatkowych polegający na zwolnieniach od podatku dochodowego cechuje się wysoką efektywnością i minimalnym ryzykiem po stronie państwa, ponieważ mogą z niego korzystać jedynie te podmioty gospodarcze, które faktycznie realizują inwestycje gospodarcze i osiągają przy tym zyski. Przez dwudziestokilkuletni okres działania ustawy o SSE nie dostosowano jednak instrumentu ulg do zmieniających się potrzeb i wyzwań ekonomicznych. Dopiero niniejszy projekt jest próbą dostosowania tych narzędzi zachęt do nowej rzeczywistości gospodarczej. Instrument zwolnień podatkowych dostępny będzie w wypadku nowych inwestycji, które według polskiego ustawodawstwa oraz zgodnie z definicją Komisji Europejskiej obejmują utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje, przy czym dotyczy to inwestycji spełniających kryteria ilościowe, nakłady inwestycyjne, i kryteria jakościowe zgodne ze strategią odpowiedzialnego rozwoju, weryfikujące wpływ inwestycji na rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wpływ na rozwój regionu. W projekcie ustawy proponuje się, biorąc pod uwagę zdiagnozowane problemy na tym polu, wprowadzenie następujących rozwiązań: po pierwsze, całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów; po drugie, wyznaczenie okresu korzystania ze zwolnienia podatkowego; po trzecie, wzmocnienie roli spółek zarządzających w systemie obsługi inwestora i, po czwarte, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zgodnie z SOR.

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, biorąc pod uwagę wszystkie powyższe walory tej regulacji, pozytywnie opiniuje projekt zawarty w druku poselskim nr 2307 i rekomenduje skierowanie tego projektu do pracy w komisji sejmowej. Głos teraz zabierze pani poseł Mirosława Nykiel z klubu Platforma Obywatelska. Pani Minister! No, pan premier Morawiecki na kongresie ekonomicznym w Krynicy zapowiedział bardzo szumnie: Polska jedną strefą ekonomiczną. Później to zostało potwierdzone przyjętą ustawą. Ale od tamtej pory tak naprawdę nic się nie zmieniło. Dzisiaj mamy projekt ustawy, która pozwala na takie alternatywne inwestycje w stosunku do tych realizowanych w ramach obecnie działających specjalnych stref ekonomicznych, czyli inwestycji opartych o ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych. I ja się bardzo ucieszyłam, bo niejednokrotnie zwracałam uwagę też na ten długi proces zmiany granic poszczególnych stref ekonomicznych i dostosowywania się do długotrwałego procesu działania inwestorów. I na tym moja radość się skończyła, bo popatrzyłam do projektu ustawy i tam kompletnie o tym nic nie wiadomo, bo tak naprawdę najważniejsza rzecz, jaka jest, to clou tej ustawy, to jest właśnie ten cały system zwolnień podatkowych uzależnionych od kryteriów jakościowych, a o tym niewiele jest w ustawie, dopiero to będzie w rozporządzeniu. Dlatego tutaj ta moja radość nie trwała długo. Tak samo jak rozmawiam z przedsiębiorcami, dopytują, kiedy rozporządzenie, które będzie określało, w jaki sposób cały system zwolnień podatkowych dla inwestorów będzie na jakim etapie procedowania tej ustawy. Dzisiaj tak naprawdę trudno mi się odnieść, bo intencje są dobre, ale jak wiemy, nasze porzekadło mówi, że dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane.

Mam nadzieję, że to nie będzie tylko takie, jak jest teraz w ustawie zaprojektowane, że te rady mogą powstać, ale nie muszą powstać, nie ma obliga. Jest obligo? Nie ma, jeśli chodzi o te rady.

Czy państwo im pozwolicie na takie bardziej arbitralne podejście, czy też państwo z góry będziecie narzucać to, co oni mają osiągnąć, bo w jaki sposób te cele zakładane w ustawie możecie, musicie uzyskać? I wielu ekspertów też, może nie tak wielu, ale przynajmniej z kilkoma rozmawiałam, ma wątpliwość, czy właśnie ten projekt ustawy nie spowoduje odwrotnego skutku do zakładanych celów. Bo jeśli jednostki samorządu terytorialnego i te spółki zarządzające będą miały dużą swobodę, to moim zdaniem będzie im bardziej zależało na tym, żeby przyciągnąć ten strumień inwestycji, coraz większy. Tymi kryteriami bardziej ilościowymi będą się kierować, miejscami pracy, a nie będą się za bardzo przejmować, że to jest całościowo jakoś niezrównoważone, i nie będą się przejmować tym, że tam jest dużo powiatów w danym regionie. Tutaj rząd ma inne cele, czyli chodzi o tę spójność celów i możliwość realizacji przez te spółki. Jakie im przyświecają przesłanki? Oni biorą przede wszystkim położenie, infrastrukturę, zasoby pracy, jakość życia. Co tam jeszcze biorą? Jeśli będą mieć możliwość wyboru w całej Polsce, to sobie wybiorą dowolnie, a niekoniecznie tam, gdzie państwo chcecie, na danym terytorium, bo tam trzeba zrównoważyć. Jesteśmy jako klub za skierowaniem procedowanej ustawy do dalszych prac w komisji, ale pod warunkiem, że na etapie prac sejmowych zostanie przedstawione rozporządzenie, które jest clou tego projektu. Wysoka Izbo! Kukiz’15 murem stoi za polskimi przedsiębiorcami, a także tak samo za pracownikami, dlatego uważamy, że Polska rzeczywiście powinna być jedną wielką strefą ekonomiczną, która będzie wspierała wszystkich, którzy inwestują na terenie Polski, wszystkich przedsiębiorców, a w szczególności te małe, średnie i mikrofirmy, bo to one najczęściej mają 100-procentowo polski kapitał i to na nich w 70% opiera się nasza gospodarka. Tym małym podmiotom też trudniej konkurować z wielkimi międzynarodowymi koncernami, które, jak wiemy, nieraz dostają dotacje rządowe, tak jak Mercedes - 81 mln, JP Morgan ostatnio - 20 mln zł. Niestety te największe firmy też najczęściej unikają płacenia podatków. Dlatego skierowanie tego projektu w szczególności do tych małych, mikro- i średnich przedsiębiorców jest bardzo ważne. Uważamy, że ta ustawa tworząca jedną wielką strefę ekonomiczną powinna być przyjęta w rzeczywistości już kilka lat temu. Dlatego mamy nadzieję, że wejdzie ona w życie możliwie jak najszybciej. Mam jeszcze pytania dotyczące rozporządzeń, m.in. o maksymalną intensywność regionalnej pomocy. Tam występuje dosyć duże zróżnicowanie pomocowe, jeżeli chodzi o województwa. Tylko problem jest taki, że w tych bogatszych województwach są też biedniejsze powiaty i wygląda na to, że te biedniejsze powiaty w bogatszych województwach stracą, a może bogatsze w tych biedniejszych dzięki temu zyskają, pomimo że województwa, jak wiemy, ze sobą graniczą i może to doprowadzać do pewnego zachwiania tego systemu. Kolejna kwestia, z tego, co widziałem, to tereny tych powiatów, które nie są też spójne terytorialnie, czyli te strefy ekonomiczne to nie jest po prostu obszar, który da się wyrysować jedną kreską, tylko one się przenikają między sobą, nie wiem, z jakich powodów.

Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Nowoczesna co do rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, druk nr 2307. Rzeczywiście jest to realizacja planu pana premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział, że chciałby potraktować Polskę jako jedną strefę ekonomiczną. Proponowany w ustawie mechanizm wsparcia ma zastąpić tak na dobrą sprawę specjalne strefy ekonomiczne, które przestaną funkcjonować w 2026 r. Ustawa wprowadza pojęcie nowej inwestycji, czyli takiej, która jest związana z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie. Wysokość wsparcia i minimalna wielkość inwestycji zależne są od kryteriów jakościowych - zgodność inwestycji z krajową strategią rozwoju, i ilościowych - wysokość bezrobocia w powiecie.

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, obszary, na których ustawa jest realizowana, i wyznaczy zarządzających obszarami. Podlegają oni przepisom o zasadach zarządzania mieniem Skarbu Państwa. Zarządzający mają przyciągać inwestycje, udzielać inwestorom informacji, pomagać im w kontaktach z administracją, współpracować z lokalnymi szkołami, udostępniać przedsiębiorcom mienie, którym zarządzają.

Zarządzający spośród zgłoszonych kandydatów, na podstawie oceny i wiedzy oraz doświadczenia, powołuje radę obszaru, w skład której wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, w tym mikro-, małych i średnich, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach obszaru oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego. Udział w radzie jest nieodpłatny. Decyzję o przyznaniu ulgi podejmuje minister gospodarki, na okres od 10 lat do 15 lat. Regulamin przyznawania ulgi, kryteria ilościowe i jakościowe, listę działalności, w przypadku których ulgi nie przysługują, sposób weryfikacji kryteriów, sposób ustalania wysokości wsparcia określa Rada Ministrów. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw budżetu może wstrzymać program ulg, czyli wyznaczyć okres, w jakim nie są wydawane nowe decyzje o przyznaniu ulgi. Warunki, jakie musi spełniać przedsiębiorca, rodzaj inwestycji, zatrudnienie, wysokość kosztów kwalifikowanych i wysokość wsparcia ustala się indywidualnie. Decyzja o przyznaniu wsparcia może zostać uchylona, jeśli przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności lub nie spełnia warunków udzielenia wsparcia, albo na wniosek samego przedsiębiorcy. Wówczas przedsiębiorca musi zwrócić otrzymaną pomoc. Urzędnicy ministra prowadzą kontrole cykliczne i doraźne spełniania tych warunków. Zdaniem autorów ustawy możliwość uzyskania wsparcia inwestycji na terenie całego kraju jest główną zaletą programów inwestycyjnych u naszych sąsiadów, w Czechach, na Węgrzech czy w Słowacji. W odróżnieniu od specjalnych stref ekonomicznych proponowany system w znacznie większym stopniu wspiera inwestycje sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych nie jest uchylona, więc będą funkcjonować tak na dobrą sprawę dwa systemy równoległe. Faktem jest, że ta ustawa określa tak z grubsza zasady funkcjonowania tych obszarów, natomiast nie będę ukrywał, że zawsze diabeł tkwi w szczegółach i będziemy czekać na rozporządzenia, które dokładnie doprecyzują, jak to ma rzeczywiście wyglądać.

Generalnie jesteśmy za tą ustawą. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Mieczysława Kasprzaka z Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów. Pani Minister! Wysoka Izbo!

Nie było lepszego rozwiązania do tej pory i trzeba oddać cześć i honor tym, którzy pracowali nad tym przez lata, udoskonalali te rozwiązania, zamiast stwierdzać politycznie: my mamy w tej chwili idealne rozwiązanie.

Potrzebne są zmiany, oczywiście, trzeba to doskonalić, poprawiać, ale nie widzę tutaj jakiejś rewolucji, bo to zależy od przedsiębiorców, zależy od szeregu innych spraw, które decydują o tym, czy będzie kapitał, czy będzie chęć inwestowania, czy przyjdą przedsiębiorcy i czy to, czy inne miejsce im się spodoba.

Natomiast powiem tak: sama nazwa i samo takie wizerunkowe głoszenie: Polska jedną wielką strefą niczego jeszcze nie zmienia.

Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do dyskusji. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu. Przepraszam.

Po pierwszym pytaniu zamykam listę. Wysoka Izbo! Wiele obszarów kraju o sporej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w rzeczywistości nie posiada wolnych zasobów ludzkich.

Moje pierwsze pytanie: Skąd takie dane i czy są one realne? Przedsiębiorcy obawiają się, że skutki zawyżonych oczekiwań co do nowych miejsc pracy, które nie będą w stanie powstać, będą przerzucane właśnie na nich. To będzie grozić nawet zwrotem całości umorzonego podatku w okresie zwolnienia. Uzależnienie zwolnienia podatkowego od oczekiwań co do nowych miejsc pracy będzie hamować nowe inwestycje. Poza tym małe firmy raczej nie spełnią kryteriów ilościowych zależnych od stopy bezrobocia w miejscu inwestycji, mimo iż zostały one znacznie obniżone. Zwłaszcza kryteria jakościowe jak zatrudnienie kadry ze specjalistycznym wykształceniem, utworzenie dobrze płatnych miejsc pracy, współpraca z ośrodkami badawczymi mogą im sprawiać trudność. Pani poseł, bardzo dziękuję. Proszę o zadanie pytania panią poseł Mirosławę Nykiel z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Pani Marszałek! Pani minister, mam pytanie odnośnie do tego rozporządzenia, o którym mówiłam: Kiedy, na jakim etapie prac sejmowych nad projektem państwo przedstawicie te założenia jakościowe i pokażecie państwo rozporządzenie? Czy on będzie ujednolicony w całej Polsce czy państwo pozwolicie spółkom zarządzającym na bardziej arbitralne podejście? Proszę o zadanie pytania pana posła Ryszarda Wilczyńskiego z klubu Platforma Obywatelska. Pani Minister! Zdecydowanie proszę o możliwość pełnej wypowiedzi, bo będę mówił wyłącznie merytorycznie.

Natomiast jest pytanie, czy to będzie dobry instrument interwencji państwowej. Mówię do pani minister. Pytanie, czy tak będzie. W tej ustawie nie ma języka, nie ma tu filozofii ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Na dodatek jeszcze państwo de facto bajpasujecie samorządy, w szczególności samorząd województwa. Jest mowa, że te inwestycje będą delimitowane, a będzie to robił minister, te obszary będą delimitowane, ale gdzie akty zasadnicze, które mówią o rozwoju obszaru, bo przecież samorząd województwa jest predysponowany do prowadzenia polityki regionalnej i prowadzenia rozwoju na swoim obszarze. Tego tutaj nie ma. Mamy tylko taki mechanizm, że to przedsiębiorca aplikuje, pisze wniosek.

Mam pytanie odnośnie do tego rozporządzenia, bo tam są wykluczane różnego rodzaju branże. To przecież branża kreatywna, twórcza, miękka, ale z dużym potencjałem, to też różnego rodzaju animacje 3D. Przecież Polski Instytut Sztuki Filmowej dostaje co roku wielomilionowe dotacje. Nie wiem, czy jest to dobra decyzja wykluczanie właśnie tych działalności. Prosiłbym może o ponowne pochylenie się nad tą częścią. Dziękuję. Pytanie teraz zadaje pan poseł Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Co w tej chwili, po tych zmianach takiego się stanie, że przedsiębiorcy na tym terenie się pojawią, jeżeli już mieli wszystko: załatwioną sprawę ziemi, poszerzenie strefy i infrastrukturę?

Proszę o zadanie pytania pana posła Jerzego Meysztowicza z klubu Nowoczesna. Wysoka Izbo! Mam pytania, dlatego że naturalną rzeczą jest - ze względu na to, że specjalne strefy ekonomiczne zostały dobrze skomunikowane, jest tam całkiem dobra infrastruktura, bo to decydowało o tym, że tam lokowały się inwestycje - że wokół tych stref są również tereny, które mogą być atrakcyjne dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli uzyskać ulgi w ramach tej ustawy, ale nie będą już na terenie strefy.

Dziękuję bardzo.

Pani minister, czy nie brała pani pod uwagę przede wszystkim połączenia tej ustawy z planami zagospodarowania przestrzennego?

Kolejna kwestia to środki unijne, które już się kończą, a przygotowanie nowego terenu, bo mówimy o terenach pozastrefowych, wymaga dużych nakładów. W tej ustawie nie ma żadnej pomocy strefy w przygotowaniu infrastruktury. Przedtem takie możliwości były.

Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam pytanie o terytorium, o to, jak zostało ono podzielone na obszary, które mają być zarządzane przez organ zarządzający, z uwzględnieniem - jak napisano - spójności terytorialnej, powiązań gospodarczych oraz granic powiatów. W drodze rozporządzenia, którego projekt jest dołączony do druku, podzielono Polskę właśnie na takie obszary, które miały te cechy spełniać: spójność terytorialną, powiązania gospodarcze i granice powiatów. Proszę państwa, Wielkopolska, z której jestem: cztery strefy i cztery podmioty zarządzające - kostrzyńsko-słubicka, łódzka, słupska i wałbrzyska. Teren bliższy, z którego jestem, powiat pilski, jest zarządzany przez kostrzyńsko-słubicką, czarnkowsko-trzcianecką, gdzie mieszkam, które sąsiadują ze sobą przez słupską. Jakież tutaj, proszę państwa, mamy powiązania? To jest wchodzenie trochę w kompetencje samorządów bez konsultacji z marszałkami. Być może się mylę.

Proszę o zadanie pytania pana posła Krzysztofa Gadowskiego z klubu Platforma Obywatelska. Pani Marszałek! Pani Minister! Państwo w swoim projekcie mówicie, że zarządzający powołuje radę rozwoju obszarów gospodarczych.

I drugie pytanie, pani minister. Minister w programach dla Śląska np. mówi, że te tereny zostaną przekazane np. do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Czy w sensie funkcjonowania, wejścia w życie tej ustawy taka możliwość będzie, czy nie?

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo się cieszę, że dzisiaj debatujemy nad projektem ustawy, która w założeniu ma bardzo szczytne cele - wsparcie inwestycji. Natomiast mam też pewne doświadczenie z przeszłości związane z moim województwem, województwem opolskim, kiedy to województwo było dosyć długo karane nieposiadaniem żadnej strefy ekonomicznej. Dopiero po kilku latach mieliśmy okazję rozszerzyć strefy wałbrzyską czy też katowicką na podstrefy w województwie opolskim. Dzisiaj państwo, przedstawiając projekt tej ustawy, mówicie o tym, że decyzje o wsparciu będą wydawane na czas oznaczony: na 10 lat, 12 lat bądź 15 lat, w zależności od intensywności pomocy publicznej w danym województwie.

Czy one będą uzależnione od tego, jakie inwestycje się pojawiają? Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania panią poseł Zofię Czernow z klubu Platforma Obywatelska. Pani Marszałek! Pani Minister! Rozwój przedsiębiorczości jest bardzo ważny dla polskiej gospodarki i wszelkie przepisy, które się do tego przyczyniają, absolutnie zasługują nie tylko na uwagę, ale i na wsparcie. Ale chciałam zapytać o skutki. Mianowicie chodzi o dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Nie znalazłam żadnego przepisu, który by mówił o rekompensatach dla tych jednostek. Proszę powiedzieć, co z tymi dochodami.

Proszę o zadanie pytania pana posła Jana Warzechę z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Wysoki Sejmie! Pani Minister! Przedstawiony projekt odpowiada na postulaty wielu środowisk biznesowych i samorządowych, jednak proszę o doprecyzowanie, o odpowiedź na kilka pytań. Jakie narzędzia zostaną wykorzystane na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki w planowanej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” Z pomocą jakich instytucji prawnych omawiany projekt zapewni wsparcie przedsiębiorcom prowadzącym lub chcącym prowadzić działalność gospodarczą w regionach zmagających się z problemami restrukturyzacyjnymi oraz adaptacyjnymi, czyli najczęściej w małych i średnich miastach, które utraciły posiadane niegdyś funkcje społeczno-gospodarcze? Czy rząd nie obawia się, że duże aglomeracje miejskie, jak również regiony lepiej rozwinięte oraz właściwie skomunikowane z naszymi partnerami w Unii Europejskiej, głównie te z dużymi ośrodkami akademickimi, skonsumują większość korzyści powstałych w wyniku wdrożenia omawianego projektu? Pytam o to, bo jestem przekonany, że rządowi przyświeca cel, [[Dzwonek]] aby realizacja projektu: Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną nie odbyła się kosztem średnich miast, a także regionów peryferyjnych o mniejszym znaczeniu gospodarczym i stopniu rozwoju. Dziękuję. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Teraz proszę o zabranie głosu panią minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz.

Pani Marszałek! Przede wszystkim chciałam podziękować serdecznie za szczegółową, detaliczną lekturę ustawy.

Powiem jednocześnie, że ta ustawa była opracowywana naprawdę, również metodologicznie, w bardzo dobry sposób, tzn. pracowaliśmy zarówno z zarządami spółek strefowych, jak i z przedsiębiorcami - z tymi, którzy już dzisiaj korzystają z tych przywilejów strefowych, jak i z potencjalnymi - jak również z samorządami, panie pośle.

To na pewno wejdzie w życie równo z ustawą, nie będzie tutaj żadnego opóźnienia. Zachęcam państwa do lektury. Kryteria jakościowe, które tam przyjmujemy, są podzielone na cztery kategorie uwzględniające rozwój strukturalny, rozwój naukowy, zrównoważony rozwój, rozwój zasobów ludzkich. Minimalne kryteria wejścia to uzyskanie 6 punktów, przy czym obniżono to do 5 punktów dla obszarów z intensywnością pomocy publicznej do 35% i do 4 punktów - z intensywnością pomocy publicznej, która może być 50-procentowa. Wśród tych kryteriów jakościowych, jakie wymieniliśmy, jest utworzenie przez inwestora centrum badawczo-rozwojowego czy utworzenie centrum usług wspólnych.

Następna wątpliwość zgłoszona w wystąpieniu to to, czy nie obawiamy się tego, że przedsiębiorcy nie wybiorą tych najlepszych, i tak atrakcyjnych miejsc. Jeżeli mówimy o mapie pomocy publicznej, to ona sama w sobie w pewnym stopniu te ograniczenia tworzy.

On istotnie ma przyciągnąć ich w te miejsca, gdzie ta pomoc publiczna jest i tak oferowana.

W wystąpieniu pana posła Meysztowicza, jak rozumiem, popierającego ideę nowej ustawy strefowej, pojawiło się odwołanie do Czech i do Słowacji. Kiedy prezentowaliśmy w ogóle założenia do ustawy, wskazywaliśmy właśnie na te dwa modele takiego dynamicznego udzielania pomocy publicznej w zależności od zapotrzebowania inwestorów.

Odpowiadając na uwagę pana posła Kasprzaka, muszę powiedzieć, że modestia, a zatem pokora, jest tą cnotą, którą staram się kierować w swojej pracy codziennie i każdego dnia. Powiedziałam tylko, że wyczerpał się model, dlatego zajęliśmy się przygotowaniem nowego, doceniając to, co w strefach się działo.

Poza tym wielokrotnie wspominałam - myślę, że jest to praktyka, o której możemy sobie tutaj ponad podziałami politycznymi jasno powiedzieć - że bardzo często instrument strefowy był wykorzystywany, zwłaszcza w pewnych sekwencjach przedwyborczych, jako pewien instrument dodatkowo wzmacniający bądź osłabiający kampanie wyborcze i ochoczo włączano do terenów strefowych tereny zalewowe, tereny pod dużą trakcją elektryczną.

A zatem te tereny są nadal terenami inwestycyjnymi, nowa ustawa ich nie wyłącza, one nadal będą mogły być oferowane, natomiast siłą nie zmusimy nikogo do tego, aby na tych terenach się pojawił.

Myślę, że ta ustawa jest właśnie wprost przede wszystkim realizacją założeń polityki rozwojowej wpisaną w „Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”

Odwołując się do kolejnego pytania, dotyczącego troski o ubytek we wypływach z podatku, które byłyby wyższe, gdyby teren nie został objęty strefą, chcę powiedzieć, że mówimy o tym, że gdyby tego przywileju nie było, danej inwestycji nie byłoby w ogóle.

Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, zawarty w druku nr 2307, do Komisji Gospodarki i Rozwoju w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Po zakończeniu dyskusji Sejm omyłkowo skierował ten projekt niezgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu. Propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu jest skierowanie tego projektu do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm tę propozycję przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 2160 i 2340) Proszę pana posła Waldemara Budę o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzyła przedmiotowy projekt na posiedzeniach w dniach 6 lutego oraz 19 marca 2018 r.

Chodzi o sytuacje takie, jak opłata od pozwu o roszczenie majątkowe z tytułu zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennej lub zbrodni agresji, oraz ujęte w ust. 1d:

Podsumowując, komisja wnosi o uchwalenie projektu według treści wynikającej ze sprawozdania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest kontynuacją nowelizacji ustawy o IPN-ie, którą niedawno Sejm przyjął. Ta ustawa o IPN-ie wywołała burzę, jak państwo wiecie. Wywołała też oświadczenia sekretarza stanu USA o zagrożeniu strategicznego partnerstwa z Polską. Kongres amerykański, zamiast zajmować się naszymi wnioskami o to, żeby obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce z rotacyjnej przekształcić w stałą, zajmuje się teraz ustawą o IPN-ie. Komitet Żydów Amerykańskich, organizacja bardzo zasłużona w lobbowaniu na rzecz wejścia Polski, przyjęcia Polski do NATO - lobbowała za tym bez żadnych warunków dotyczących, nie wiem, reprywatyzacji czy czegoś innego - organizacja, która pomaga nam zwalczać używanie sformułowania polskie obozy śmierci, która niedawno otworzyła biuro w Warszawie, wyraził ubolewanie z powodu tej ustawy. Stosunki z Izraelem, które rozwinęły się bardzo dobrze - i z diasporą żydowską i jeśli chodzi o dialog polsko-żydowski, który pozwala nam przedstawiać Polskę jako miejsce, gdzie Żydzi przez wiele setek lat mieli schronienie - w tej chwili uległy gwałtownemu zepsuciu, bo Polska jest podejrzana po tej ustawie o IPN-ie o to, że chce w jakiś sposób ograniczać dyskusję nad Holocaustem, że ocaleni z Holocaustu czy ich dzieci będą musieli się tłumaczyć ze sformułowań zawartych w pamiętnikach, gdzie coś jest niepochlebnego o Polsce czy coś złego. Trzeba będzie udowadniać przed sądem, że to są fakty, bo inaczej grożą za to 3 lata więzienia. Dialog z Izraelem również jest z powodu tej ustawy niezwykle zepsuty, jak i te wszystkie osiągnięcia, które mieliśmy przez ostatnie lata w tej dziedzinie. Również jest kwestia dialogu historycznego z Ukrainą, który się dobrze rozwijał, wielkim wysiłkiem duchownych po obu stronach, Jana Pawła II, który o tym mówił, poprzednich prezydentów Polski i prezydentów Ukrainy, którzy wydawali w tej sprawie wspólne oświadczenia czy wspólnie uczcili ofiary cywilne po obu stronach.

Już nie mówię o opinii polskich historyków - od Sławomira Cenckiewicza do Andrzeja Friszkego - którzy protestują przeciwko tej ustawie. Ale to wszystko, proszę państwa, PiS-owi jest za mało, to jeszcze jest za mało. Do tej burzy, która się toczy wokół tej ustawy, PiS postanowił dolać jeszcze benzyny, do tego ognia, do tego pożaru i zgasić go za pomocą benzyny. Ta ustawa, którą dzisiaj rozpatrujemy, dotyczy zniesienia opłat za pozwy wynikające z ustawy o IPN-ie wnoszone przez organizacje, które mają wpisane w statucie zadanie obrony dobrego imienia narodu polskiego czy Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym te organizacje. Ta opłata teraz wynosi 5%, ona ma na celu pokrycie kosztów sądowych, ma również pewne znaczenie dyscyplinujące, że nie wnosi się pozwów w sprawach absurdalnych, nie wnosi się pozwów o odszkodowania z jakimiś horrendalnymi kwotami. Teraz państwo chcecie znieść tę dyscyplinę i każda organizacja, która ma to zapisane w statucie, będzie mogła wnosić sprawy przeciwko każdemu. Jeśli ktoś np. powie: Zastanawiam się, czy Polakami da się rządzić bez bata. Drugi cytat tego samego autora: Wytworzyłem całe mnóstwo pięknych słówek, które naród polski stawiają w rzędzie idiotów - to mówił Józef Piłsudski. Inny cytat, który wszystkim państwu chyba jest znany: Polsko, pawiem narodów byłaś i papugą, a teraz jesteś służebnicą cudzą - Słowacki.

Otóż jeśli jakaś organizacja uzna, że ktoś, kto powtarza takie słowa czy tego typu sformułowań dzisiaj używa, obraża naród polski i jego dobre imię, będzie mógł wystąpić z nieograniczonym pozwem na nieograniczoną kwotę. Chodzi również o obecne sformułowania dotyczące Polaków dzisiaj. Dlatego, proszę państwa, Platforma Obywatelska będzie głosować przeciwko tej ustawie, bo zwolnienia z kosztów, jeśli to są kombatanci czy ofiary zbrodni wojennych, można zawsze uzyskać w sądzie indywidualnie. Dziękuję, panie pośle. Nie ma pana posła. Proszę o zabranie głosu panią poseł Kornelię Wróblewską z klubu Nowoczesna. Wysoka Izbo! Ta ustawa to nic innego jak dalszy ciąg sagi pn. „Niepotrzebna i zła ustawa o IPN” W słynnej ustawie skrytykowanej już chyba przez wszystkich wprowadziliście oprócz znanych wszystkim przepisów karnych przepisy umożliwiające dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkalowanie narodu polskiego. Z takim pozwem mogą wystąpić również organizacje społeczne. I teraz, by ułatwić osobom zainteresowanym wytaczanie takich spraw, zwalniacie je, jak również kombatantów i ich dzieci, z opłaty za złożenie takiego pozwu. Szanowni państwo, takie działanie mija się z celem. Wiem, że chcecie, by takich pozwów było jak najwięcej i żeby wszyscy niewygodni musieli stanąć przed sądem i tłumaczyć się, że nie ma podstaw do żądania od nich np. 10 mln zł za jakieś słowa rzucane tak naprawdę nie przeciwko państwu polskiemu, a przeciwko aktualnej władzy. Dlaczego mieszacie w to kombatantów? Dlaczego dajecie ten przywilej ich zstępnym?

To jest sprzeczne z zasadą równością obywateli, gdyż segreguje się ludzi na tych bardziej uprzywilejowanych, czyli mających w swym rodzinnym otoczeniu kombatanta, i na tych, którzy takiego kombatanta w swojej rodzinie nie mają. Po pierwsze, mamy tu do czynienia z przedmiotowym traktowaniem osób najbardziej zasłużonych dla naszego narodu. Po drugie, to wszystko budzi poważne wątpliwości konstytucyjne związane z naruszeniem lub wręcz złamaniem konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. Prowadząc politykę historyczną zamiast polityki przyszłości i rozwoju, dążycie do skłócenia obywateli ze sobą w ramach jednego państwa. Nasza ojczyzna? W jaki sposób? Zyska na tym tylko władza. Wyciągacie trudne sprawy i rozdrapujecie dawno zabliźnione rany, dając tym samym przyzwolenie nowym pokoleniom na wzniecanie wojny polsko-polskiej, na ocenianie, kto jest lepszym, kto gorszym sortem Polaków. Zainwestujecie we wnoszone procesy, bo gdy będą zwolnione z opłat, to zapewne będzie ich sporo, a koszty będzie musiało ponieść w takiej sytuacji państwo polskie. Ewentualną wygraną przekierujecie na cele własnej działalności izolującej Polskę na arenie międzynarodowej, na hojne premie uznaniowe, tabuny niedoświadczonych asystentów i takie biznesy jak SKOK Holding czy spółka Srebrna, dla niepoznaki prowadzone poza granicami państwa. Takie działania nie tylko nie zamkną ust obywatelom, ale dodatkowo jeszcze znacząco przedłużą postępowania, w szczególności w dużych miastach. Ta ustawa, zwalniająca z jakichkolwiek opłat, a opłaty, przypomnę, służą powstrzymaniu przed nieuzasadnionymi pozwami, spowoduje, że będzie można żądać milionowych odszkodowań, nie płacąc nic, a sędziowie będą musieli rozpatrywać każdą sprawę i zapewne najczęściej oddalać powództwa. Każdą, bo proponowana ustawa zakłada, że w tym temacie nie ma spraw nieuzasadnionych. Niestety jest to błędna logika, szanowni państwo. Efekt? Dopóki sytuacja się nie unormuje, w największych sądach zatory w rozpatrywaniu spraw wzrosną do poziomu utrudniającego normalne działanie organu, a zatem podważą skuteczność sądów, pozbawiając obywateli szans na załatwienie ważnych dla nich osobiście kwestii. Ta ustawa jest nie do przyjęcia w takiej formie. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Paszyka, Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Chciałbym w imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem projektowanej nowelizacji jest rozszerzenie katalogu pism, które nie podlegają opłacie, o pozwy w sprawach roszczeń majątkowych o ochronę dóbr osobistych. Nowe przepisy obejmą kombatantów, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i ich zstępnych.

Obecnie takie powództwa są objęte ogólną zasadą, zgodnie z którą opłata od ich skutecznego wniesienia wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Wysoka Izbo! Prawo do dochodzenia przed sądem ochrony dóbr osobistych jest jednym z ważniejszych przysługujących nam praw. Opłaty za pozwy mają jednak swój konkretny cel. Celem jest odsianie osób, które zalałyby sądy niezliczoną ilością pozwów, oskarżając każdego wokół o naruszenie ich dóbr. Wszyscy wiemy, że istnieje kategoria osób nad wyraz wrażliwych na swym punkcie. Istnieje też kategoria organizacji chcących pozwać cały świat za to, że nie podziela określonej wersji historii. Musimy pamiętać, że postępujące ograniczenie stosowania opłat może doprowadzić do niekontrolowanego przyrostu spraw w sądach i w efekcie jeszcze bardziej spowolnić ich działanie. Należy też zauważyć, że brzmienie projektu nie pozwala precyzyjnie określić, komu będzie przysługiwało zwolnienie i co oznacza słowo „ofiara” Nie ma w projekcie zdefiniowanego pojęcia „ofiara” Rodzi to określone trudności interpretacyjne i może utrudnić stosowanie przepisów ustawy. Zwraca też uwagę to, że autorzy projektu nie podają spodziewanych kosztów wprowadzenia projektu, nie mówią nam, jakie będą skutki finansowe wejścia w życie tych przepisów. Wysoka Izbo! Niewątpliwie powinno nam wszystkim zależeć na ochronie dobrego imienia kombatantów - tu należy zrobić ukłon w stronę projektodawców - tak samo jak na ochronie wizerunku Polski i narodu polskiego.

Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów niestety nie widzi możliwości poparcia projektu w tym kształcie. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Stanisława Piotrowicza z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kiedy wsłuchuję się w wystąpienia moich przedmówców, wydaje mi się zasadne przytoczenie roty ślubowania poselskiego: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” Wydaje się zasadne zwrócić uwagę na polską rację stanu. Polską racją stanu jest służyć wiernie Rzeczypospolitej i narodowi polskiemu, i to ślubowali wszyscy posłowie. Obrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej winna głęboko leżeć na sercu każdemu posłowi. Trzeba wrócić do tekstu ustawy, bo wkradają się pewien chaos i nieporozumienie: nie pobiera się opłat od pozwu o ochronę dóbr osobistych od kombatantów, a więc od tych ludzi, którzy w sposób szczególny zasłużyli się Rzeczypospolitej Polskiej. W innych przepisach gwarantujemy kombatantom wsparcie, ochronę, szacunek dla ich wkładu w walkę o dobro Rzeczypospolitej, o jej suwerenność i niepodległość, a teraz rozdzieramy szaty - mówię tu o posłach opozycyjnych - że oto zostaną oni zwolnieni z opłaty sądowej, i podnosi się kwestię nierównego traktowania podmiotów. Tu nie chodzi o pozwy kombatantów w ich sprawach prywatnych, majątkowych. Albo zła wola, albo manipulacja, albo nieznajomość tekstu ustawy skłaniała do takich wystąpień, jakich świadkami byliśmy przed chwilą. Otóż mamy wąsko ograniczony zakres przedmiotowy tych pozwów i warto, ażeby to w tej Izbie wybrzmiało. Te pozwy dotyczą ochrony dóbr osobistych, gdy sprawa - wyraźnie jest powiedziane - dotyczy patriotycznych tradycji zmagań narodu polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem. Zwolnienie z opłaty sądowej kombatantów. Kombatanci zazwyczaj są w dość trudnej sytuacji materialnej, bo takie są realia. Dostęp do sądu nie oznacza, że można przyjść do sądu, ale dostęp do sądu oznacza, że można się domagać skutecznie rozstrzygnięcia wniesionej sprawy, że można się domagać rozstrzygnięcia wniesionej sprawy. Wysoka opłata sądowa dla tych ludzi często jest barierą uniemożliwiającą dostęp do sądu. A więc mamy tutaj do czynienia ze zwolnieniem przedmiotowym - kombatantów i podmiotowym - ściśle określonej kategorii spraw. Również dziwię się, że państwo tak wielokrotnie podkreślacie znaczenie organizacji pozarządowych w różnych kwestiach, a nie chcecie dostrzec możliwego wkładu tych organizacji w ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej. Przecież to są nasi sojusznicy. To nasz wspólny interes, to nasz poselski obowiązek. Jednocześnie pozwolę sobie złożyć w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość poprawkę zmierzającą do skreślenia z ustawy pkt 1d. Klub Prawa i Sprawiedliwości w pełni popiera projekt ustawy wraz z poprawką, którą przedłożyłem na ręce marszałka. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do zadawania pytań.

Wysoka Izbo! W niniejszej zmianie ustawy bronimy kombatantów i chcemy im dać pewien przywilej, ale mowa jest również o zstępnych i spadkobiercach. Czy posłowie wnioskodawcy tego projektu zauważyli, że rodzi to swoistą nierówność obywateli wobec konstytucji? Jak można zauważyć, zmiana ustawy powołuje kategorię Polaków, którzy mają wśród swoich przodków kombatantów, dlatego przysługuje im ważny przywilej. To nierówne traktowanie Polaków. Kolejna sprawa. Schorowani i słabi kombatanci, bo to na ogół obywatele powyżej 80. roku życia, mają do pomocy różnego typu organizacje w występowaniu do sądu z roszczeniami. Dlatego chciałam zapytać o opłatę. Czy jej likwidacja lub obniżenie nie wywoła [[Dzwonek]] takiego skutku, że będą pozwy o niebotyczne kwoty bez żadnych konsekwencji wnoszone przez organizacje? Proszę o zadanie pytania panią poseł Katarzynę Osos z klubu Platforma Obywatelska. W takim razie proszę o zadanie pytania panią poseł Zofię Czernow z Platformy Obywatelskiej. Panie Ministrze! Moja wypowiedź nie dotyczy kombatantów, bo tutaj nie mam żadnych wątpliwości i, myślę, nikt z nas nie ma wątpliwości, i sądzę, że niepotrzebnie pan przewodniczący Piotrowicz przekonywał, że jest inaczej. Słuchając wypowiedzi pana przewodniczącego, mam takie nieodparte wrażenie. Z tej wypowiedzi wynika, że to wszystko jest tak jasne i oczywiste, a już tyle poprawek do tego jednego artykułu. Przecież w komisji były poprawki, o IPN-ie mówiliśmy, że to jest błąd, i dzisiaj pan przewodniczący poprawkę składa, żeby to wykreślić. Tak że to nie jest takie oczywiste. Mam pytanie takie. Czy wnioskodawcy nie obawiają się ogromnej liczby procesów na koszt Skarbu Państwa? Bo w obecnej sytuacji w Polsce każdemu niemalże można zarzucić, [[Dzwonek]] że negatywnie wypowiada się na temat wizerunku lub pisze odpowiednie sformułowania. Proszę o zadanie pytania pana posła Marcina Święcickiego z klubu Platforma Obywatelska.

Pani Marszałek! Rozumiem, że poprawka, którą zgłosił tutaj pan poseł, zmierza do usunięcia części tych idiotycznych rozwiązań w tej ustawie, ale bynajmniej nie wszystkich. Dlatego mam pytanie do państwa: Czy gdzieś jest jakiś cywilizowany kraj, który daje takie uprawnienia, jakie państwo tutaj dajecie kombatantom i osobom zstępnym oraz organizacjom pozarządowym, żeby można było skarżyć na całym świecie, wysuwać pozwy i żeby one były zwolnione od opłat? Jeszcze raz chciałem podkreślić, że obecne przepisy pozwalają zwalniać kombatantów, jeśli nie stać ich na wniesienie tego rodzaju sprawy. Natomiast robienie jakiejś osobnej kategorii obywateli ze zstępnych kombatantów. Gdzie, w jakich krajach występują tego rodzaju rozwiązania? To raczej przypomina Turcję i Rosję, a nie jakieś cywilizowane kraje, które miałyby.

Proszę teraz o zadanie pytania pana posła Jerzego Meysztowicza z klubu Nowoczesna. Wysoka Izbo! Ja nie wiem, dlaczego. Panie ministrze, pytanie: Czy obecne przepisy nie pozwalają na zwolnienie z opłat osób, które są w trudniej sytuacji finansowej? Pozwalają. Natomiast te opłaty mogą skutkować tym, że nie będzie chorych żądań, bo jeżeli ktoś nie będzie wpłacał żadnych opłat, to zażąda milionowych odszkodowań.

O tym już pan zapomniał powiedzieć, natomiast poucza mnie pan, jak ja mam traktować swoje ślubowanie poselskie. Pan jest ostatnią osobą, która ma prawo o tym mówić, pan. Komunistyczny prokurator nie będzie mi mówił, jak ja mam się zachowywać w stosunku do polskiej racji stanu. Proszę o zadanie pytania panią poseł Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską z klubu Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo!

Natomiast bardzo proszę posłów wnioskodawców o odpowiedź na pytanie, czemu tak naprawdę służą zapisy dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Oczywiście można. To jest pytanie retoryczne, więc odpowiedź jest oczywista.

I też zawsze można by było zadać sobie pytanie, czy osoby ubogie nie mogłyby poprzestać na tym, że można by zwalniać od kosztów.

Drugie pytanie: Czy konieczność uiszczenia opłaty sądowej nie zabezpiecza w odpowiedni sposób przed wnoszeniem bezzasadnych powództw, czy właśnie takim projektem nie otwieramy, Wysoka Izba nie otwiera zbyt szeroko furtki dla wnoszenia pozwów niekoniecznie uzasadnionych? Otóż zwolnienie od kosztów sądowych, zwłaszcza częściowe, bo takim jest zwolnienie od opłaty od pozwu, nie jest instytucją, która otwiera drzwi sądów na bezzasadne roszczenia, ponieważ to jest tylko pewien element kosztów, które każdy jest obowiązany ponieść w procesie, zwłaszcza przy częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych w postaci opłaty od pozwu. Są inne opłaty, i o tym toczyła się wczoraj na posiedzeniu komisji dyskusja, dotyczące choćby należności biegłych, są opłaty od środków odwoławczych, są różnego rodzaju inne opłaty wchodzące w zakres kosztów sądowych i są wreszcie koszty zastępstwa procesowego, koszty adwokackie czy radcowskie. W związku z tym samo istnienie zwolnienia od opłaty od pozwu nie oznacza, że osoba bezzasadnie wytaczająca tego rodzaju powództwa może nie liczyć się... a właściwie ona powinna się liczyć z koniecznością zapłaty, bo bezzasadne powództwo oznacza, po pierwsze, że ponosi się koszty inne niż opłata od pozwu, po drugie, że trzeba zapłacić przeciwnikowi procesowemu w wypadku oddalenia powództwa niebagatelnej wysokości koszty adwokackie czy radcowskie. Zatem nie dyskutujemy tutaj o bezzasadnym otwieraniu drzwi do sądów, tylko o pewnej opłacie, pewnym ułatwieniu w określonej kategorii spraw ze względów społecznych, wydaje się, jak najbardziej uzasadnionych. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie?

Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! W moim oświadczeniu poselskim chciałbym przypomnieć historię rozpoczynającej obecnie swoje istnienie i funkcjonowanie nowej inwestycji realizowanej przez 30 lat z budżetu państwa, jaką jest zapora i zbiornik wodny w Świnnej Porębie. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny sezon nad Jeziorem Mucharskim, bo o nim mowa, będzie już dostępny dla wędkarzy, a na zalewie pojawią się pierwsze patrole wodne WOPR. Myślę, że dziś w początkowym momencie funkcjonowania tej pięknej, wspaniałej i okazałej inwestycji warto choć w kilku zdaniach wspomnieć historię jej realizacji, a także cenę, która nigdy nie była oszacowana, jaką musieli zapłacić mieszkańcy strefy zalewowej i obszarów przyległych do linii brzegowej obecnego zalewu. W momencie rozpoczęcia pierwszych prac zlikwidowano tam istniejące zakłady produkcyjne i inne miejsca pracy. Zakazano też wszelkich inwestycji w jakąkolwiek infrastrukturę, znacznie obniżając poziom i komfort życia mieszkańców, pozbawiając ich tym samym możliwości rozwoju i podejmowania własnych inicjatyw. Wielu z nich przez te lata musiało żyć i mieszkać na wielkim placu budowy, aby ostatecznie opuścić swoje domy i rozpocząć swoje życie na wyznaczonych terenach. Drodzy Państwo! Nie zamierzam mówić o dramacie, bo chcę mówić o sukcesie. Wracając do meritum, przypomnę, że inwestycja ta rozpoczęła się w 1986 r. i do roku 1999 była finansowana z budżetu państwa. Od roku 2004, przepraszam, od roku 2000 do roku 2004 na mocy decyzji parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej była finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co było finansowaniem nie tylko niewystarczającym, ale też chaotycznym i niekompatybilnym z rzeczywistymi potrzebami. To nie dawało ani nadziei, ani szansy na realizację tego zadania.

Określono w nim cztery kluczowe zadania, tj. budowę zbiornika, odbudowę dróg, przeniesienie linii kolejowej i ochronę zlewni, oraz wiele innych niedookreślonych inwestycji: odtworzenie budynku domu dziecka, odbudowę zabytkowego dworku w Dąbrówce, budowę lokali socjalnych dla wysiedlonych mieszkańców, odbudowę boisk sportowych i wiele innych strategicznych zadań. Pomimo w mojej ocenie świetnie wówczas opracowanego programu, brak stabilnego finansowania, wzrost kosztów pracy i materiałów budowlanych, długotrwałe procedury przetargowe, procedury wyłaniania wykonawców, a także czas trwania budowlanych procesów technologicznych wykluczyły zakończenie tej inwestycji w roku 2010. Z tych samych powodów, o których wcześniej wspomniałem, w grudniu 2013 r. Sejm wyznaczył kolejny termin na rok 2015. Był to ostatni rok finansowania tej inwestycji na mocy tego programu, ale nie był to rok jej zakończenia, bo do wykonania pozostały m.in. rozruch na mokro zapory oraz czaszy zbiornika, rozruch elektrowni, rozbiórka dróg asfaltowych i dwóch mostów, doszczelnienie galerii kontrolno-zastrzykowej na etapie piętrzenia oraz budowa dwóch lokalnych dróg. Dlatego dla zapewnienia realizacji tych zadań Sejm 13 maja 2016 r. uchwalił poselski projekt ustawy o dokończeniu budowy zbiornika w Świnnej Porębie, zabezpieczając w nim środki na realizację tych zadań. Na zakończenie dodam, że łączny koszt tej inwestycji zamyka się w kwocie 2210 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że najbliższy tegoroczny sezon nad zalewem będzie pierwszym dostępnym dla wędkarzy, turystów i amatorów sportów wodnych. Wysoka Izbo! Takie oto wydarzenia utkwiły w mojej pamięci. Postanowiłem się nimi z państwem podzielić. Zachęcam jednocześnie wszystkie panie i panów posłów do odwiedzenia tego regionu, na którego rozwój wszyscy mieliśmy wpływ. Dziękuję.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci nieodżałowanej pamięci pana Franciszka Szelwickiego. Pozwólcie państwo, że przybliżę nieco jego sylwetkę. Ukończył Technikum Mechaniczne w Świdnicy.

We wrześniu 1980 r. wstąpił do „Solidarności”

Zastaje członkiem komisji krajowej związku.

Od sierpnia 1982 r. do 1989 r. współzakłada podziemny ruch wydawniczy, jest kolporterem prasy i wydawnictw podziemnych, w tym m.in. „Tygodnika Mazowsze” oraz „Sygnałów Wojennych”

Po 1989 r. był delegatem na kolejne walne zebrania delegatów „Solidarności” regionu Śląska Opolskiego.

Cała jego działalność była przepełniona troską o dobro Polski. 23 sierpnia 2007 r. postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego pogrzeb odbędzie się w najbliższy czwartek w Lasowicach koło Otmuchowa na Opolszczyźnie. Cześć jego pamięci!

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! „Andrzejowi Zamoyskiemu, kanclerzowi wielkiemu koronnemu, w trzechsetną rocznicę urodzin” - takie motto znalazło się na stronie przedtytułowej reprintu „Zbioru praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego, który został opracowany i wydany z inicjatywy pana Jerzego Piotrowskiego, kierownika Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, dzięki finansowemu zaangażowaniu państwa Jolanty i Dariusza Grabikowskich oraz państwa Reginy i Henryka Grześkiewiczów. Ci państwo są z nami, są obecni na galerii i serdecznie ich pozdrawiamy. Andrzej Hieronim Franciszek Zamoyski herbu Jelita zapisał bogatą kartę w dziejach Rzeczypospolitej jako patriota, magnat posiadający znaczny majątek, pisarz, reformator oraz nietuzinkowy polityk. Żył w okresie wielkich wstrząsów politycznych i gospodarczych, jakie nawiedziły Rzeczpospolitą w XVIII w., nigdy nie pozostając wobec nich biernym. Urodził się 30 września 1717 r. w Gniewie jako trzeci syn Michała Zdzisława, łowczego wielkiego koronnego, wojewody lubelskiego, szóstego ordynata Zamościa oraz Anny z Działyńskich, wojewodzianki chełmińskiej. W 1742 r. dokonano podziału majątku po zmarłych rodzicach, dzięki któremu Andrzej Zamoyski otrzymał tzw. schedę drugą, obejmującą dobra bieżuńskie, kutnowskie i część beresteckich. Pozostawił po sobie w Bieżuniu wiele śladów materialnych, rozbudował rezydencję poprzez przebudowę pałacu oraz urządzenie parku z największym w Europie kanałem usytuowanym na osi założenia. Obecnie zarówno pałac, jak i jego otoczenie znajdują się w stanie agonalnym i wymagają pilnej interwencji konserwatorskiej. Trzechsetna rocznica urodzin arystokraty jest doskonałą okazją do przypomnienia jego najważniejszego dzieła, które zostało przygotowane i złożone w Sejmie w 1778 r., stanowiło projekt nowego prawa, które w rzeczywistości zawierało koncepcję gruntownej naprawy państwa. Jego pełny tytuł brzmi: „Zbior praw sądowych na mocy Konstytucyi roku 1776. przez J.W. Andrzeia Zamoyskiego, Ex-Kanclerza Koronnego, Kawalera Orderu Orła Białego, ułożony, y na Seym roku 1778. podany”, a przeszedł do historii jako „Kodeks Zamoyskiego” Kodeks Zamoyskiego” był pracą unikatową, wybitnie nowoczesną i postępową jak na owe czasy. Między innymi przejęte w znacznej mierze z postulatów ówczesnej doktryny humanitarnej przepisy likwidowały przejawy arbitralności wymiaru kary. Po odrzuceniu kodeksu przez Sejm w 1780 r. Zamoyski wycofał się z życia publicznego.

Dziękuję, pani poseł. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Aleksandra Mrówczyńskiego z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Nie widzę pana posła, zatem proszę o zabranie głosu pana posła Jacka Kurzępę z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jesteśmy, jak państwo wiecie, w reżimie działania przyjętej przez Sejm ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W ustawie był określony czas na jej wykonanie przez samorządy, a w sytuacji gdy tego nie wykonały, wojewoda, po uzyskaniu opinii IPN, może wydać zarządzenie zastępcze nadające danej ulicy nazwę zgodną z ustawą dekomunizacyjną. Rozmaicie samorządy wokół tej ustawy się organizowały, wiele wykorzystało sposobność, by zmienić historyczne i symboliczne oblicza swoich małych ojczyzn. Zbyt wiele jednak było zachowawczych, oporujących li tylko dlatego, że inicjatorem zmiany jest Prawo i Sprawiedliwość. Zdarzały się samorządy - i ich gospodarze - które mimo że same nie mają historycznie zbyt oczywistego zakorzenienia tożsamościowego w najnowszych dziejach Polski, nie chciały pójść tym tropem i na propozycje nadania zaszczytnych imion bohaterów narodowych czynów zbrojnych, nauki czy sztuki - po prostu nie skorzystały z tego. Poszły w całkowitą aksjologiczną i historyczną nijakość, rzekomo nawiązując do nazw sprzed wielu, wielu wieków bądź też idąc w stronę całkowicie nijaką, nadając nazwy: Wakacyjna, Rowerowa, Poprzeczna, Agrestowa.

Wiemy, że uczestnictwo w tego typu konsultacjach nie musi być reprezentatywne dla opinii całej społeczności, a zatem nie w tym rzecz, tylko w tym, czy chcemy, by przestrzeń symboliczna naszych miast i wsi do nas przemawiała. Jeśli tak, to w oparciu o jakie wartości i postaci? Nawiązuję w tym wystąpieniu do miasta Krosno Odrzańskie i miasta Gubin. Ziemia, która jak kania dżdżu potrzebuje zakorzenienia w tożsamości. A włodarze tych miast proponują właśnie taką totalną nijakość w nazewnictwie. Sądzę, że w większości mieszkańcy chcieliby, by bohaterami ich ulic byli giganci ducha, charakteru i niezłomności postawy, intelektu bądź niekwestionowanego dorobku twórczego.

Proszę o zabranie głosu pana posła Dariusza Bąka, klub Prawo i Sprawiedliwość.

Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda stwierdził, że chce, aby w świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości włączyli się wszyscy jego rodacy. Aby tak być mogło, należy pochylić się nad wszystkimi grupami społecznymi i uczciwie ocenić wkład w odzyskanie wolności i niepodległości. Polacy bowiem nie jeden raz wolność odzyskiwać musieli i ciężko pracować nad ocaleniem polskości. Chciałbym zatem zwrócić państwa uwagę na mieszkańców polskiej wsi. Dopóki rolnicy nie protestują, nie krzyczą o swojej krzywdzie, można się nimi nie zajmować, a nawet w majestacie prawa ograniczać ich wolność i dokładać ciężarów. Alienacja i samouwielbienie niektórych rządów pojawiają się szybko, więc trudno się temu dziwić. A ja wbrew temu uśpieniu, alienacji i krótkowzroczności pragnę przypomnieć o tym, co było na polskiej wsi i co jest dzisiaj. Tam bowiem w polskich dworach i chłopskich chatach rodziła się piękna polska kultura, która miała i ma charakter nasz - polski i uniwersalny. Wieś wydawała wielu poetów, pisarzy, uczonych wielkiego formatu, księży i polityków. Synowie wsi szli do walki, aby bronić ojczyzny i urastali do rangi narodowych bohaterów tych znanych, zapisanych przez historyków, i cichych w swojej wielkości, o których pamięta jedynie rodzina, parafia lub cała wieś. Na wsi zrodziła się solidarność między szlachtą i chłopami, widoczna we wszystkich powstaniach narodowych i w solidarności wiejskiej w czasie ucisku komunistycznego. I wreszcie tam uczono swoje dzieci szacunku do starszych, do chleba, do ziemi, bo ona jest nasza i Boża, święta. Tam żarliwie wznoszono modły do Boga, kiedy lała się polska krew i kiedy wróg usiłował wykorzenić nas z naszej tradycji. Tam zawsze znalazł się ktoś, kto skupiał wokół siebie gromadę i opowiadał starodawne dzieje, wskrzeszał bohaterski czas i uczył prawdy o świecie. Tam ksiądz przypominał, skąd rodzi się w człowieku duchowa radość i jak swoją dolę i niedolę powierzać Bogu i ojczyźnie. Tam wreszcie, na polskiej wsi inaczej niż w naszych czasach ludzie rozumieli, że prawo ludzkie, stanowione ma wyrastać z prawa Bożego i naturalnego. Człowiek o prawym, prostym sercu nie zrozumie dzisiejszego ujmowania prawa oderwanego od zasad moralnych, co sprowadza się do tego, że to, co zapisane w ustawach, ma być, choćby zagrażało życiu bezbronnych i godziło w honor ustawodawców, odczłowieczało człowieka i uczłowieczało zwierzęta. Zatem oświadczam, że te problemy są związane z piękną stroną życia polskiej wsi. Pragnę Wysokiej Izbie przypomnieć, a może też tę myśl ożywić, żeby wieś urosła do rangi naszej wspólnej sprawy, tak jak cała nasza ojczyzna, Polska. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Maciejewskiego, klub Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Człowiek jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno - tak w jednym ze swoich utworów pisał Stefan Żeromski. Dobrze byłoby, żeby każdy tak myślał, chociaż skoro nasz wielki pisarz zwraca na ten fakt uwagę, to znaczy, że z jego doświadczeń wynikało, że pozycja człowieka może być zagrożona. Czy wszystko, co tworzy, nie ma mu służyć i ułatwiać życia? Uwaga Żeromskiego wydaje się tak oczywista, że trudno z nią dyskutować. O wszystkim decyduje człowiek. Niestety także o tym, że powstają nieporozumienia i konflikty, a jak konflikty, to i ofiary tych konfliktów. Oczywiście są odpowiednie instytucje państwowe, które rozwiązują te konflikty, ale pozostaje ich skutek, czyli ból, żal, depresja powodująca wielkie zmiany w psychice ofiary i pozostająca czasem przez całe życie. Takim ludziom trzeba koniecznie pomóc, bo w obliczu przykrych i niespodziewanych zdarzeń najczęściej są bezsilni, bezradni i zrozpaczeni. Tacy ludzie nie mogą sobie znaleźć miejsca na ziemi. Tragizm tej grupy społecznej został zauważony przez państwa członkowskie Rady Europy i Unii Europejskiej, dlatego uchwalono dzień 22 lutego międzynarodowym dniem ofiar przestępstw, w którym to dniu od 1988 r. szczególnie zwracana jest uwaga na prawa ofiar.

Tę bardzo ważną dla pokrzywdzonych ludzi datę pamiętają wszystkie organizacje pozarządowe, które w swoim statucie zapisały niesienie pomocy ofiarom przemocy.

Każdy z nas może być ofiarą i właśnie dlatego istnieje ogromna potrzeba wypracowania systemu, który będzie chronił interesy przyzwoitych ludzi, który w sposób skuteczny w razie potrzeby udzieli kompleksowej pomocy, łącznie z wsparciem prawnym i psychologicznym. Tak to już w życiu jest, że póki nas problem ofiary osobiście nie dotknął, to traktujemy tę sprawę bardzo lekceważąco. Dopiero gdy sami stajemy się ofiarą, zaczynamy rozumieć, jak wiele trzeba jeszcze zrobić, by chociaż w części to, co straciliśmy w wyniku przestępstwa, odzyskać. Dopiero wtedy zauważamy, jak bardzo wiele państwo musi jeszcze zrobić, by zabezpieczyć ofierze prawa do godnego życia. Niestety administracja państwowa, co z przykrością należy stwierdzić, nie w pełni odpowiada na potrzeby ludzi pokrzywdzonych. Właśnie dlatego trzeba zauważyć, jak dużą rolę odgrywają organizacje pozarządowe, które wciąż przypominają, że ofiara potrzebuje opieki w zdecydowanie większym zakresie niż dotychczas. Dzisiaj tę opiekę zabezpieczają członkowie organizacji pozarządowych, bo są to ludzie wyjątkowo wrażliwi na krzywdę ludzką. Myślę, że niewiele się pomylę, jeśli powiem, iż tacy ludzie są nieodłącznym elementem życia osoby pokrzywdzonej, są wsparciem w walce o sprawiedliwość, o wykrycie i przykładne ukaranie winnego oraz o odzyskanie równowagi psychicznej po stracie bliskiej osoby. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzień ten minął jak każdy inny. Szkoda, że nadal w środkach masowego przekazu tak bardzo mało o nim się mówi. Właśnie w tym dniu możemy podkreślać świętość człowieka i wyrabiać, zwłaszcza u młodzieży, wrażliwość na krzywdę ludzką w możliwie szerokim znaczeniu. Sądzę, że myśląc o człowieku jak o świętości, powinniśmy traktować ją jak nakaz, którego złamać nie można nawet z najszlachetniejszych powodów, bo, jak pisał Mieczysław Wiraszko, kto w potrzebie opuszcza drugiego człowieka, wyrzeka się człowieczeństwa. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Szulowskiego, klub Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! W dniu dzisiejszym rano dotarła do mnie długo oczekiwana wiadomość. W Puławach usunięto pomnik przedstawiający dwóch żołnierzy: sowieckiego i polskiego z 1. Armii Wojska Polskiego. Potężny, wykonany z czerwonego piaskowca monument z napisem „Bohaterom wspólnych walk o wyzwolenie Puław - społeczeństwo miasta” został postawiony w 1987 r. na miejscu jeszcze większego symbolu zniewolenia, jakim był pomnik poświęcony bohaterom armii radzieckiej poległym na polu chwały. Już od dawna trwały starania środowisk patriotycznych, niepodległościowych o to, aby pomnik, potocznie nazywany pomnikiem Bolka i Lolka, zniknął z przestrzeni publicznej miasta. 30 maja 2016 r. stosowane stanowisko przyjęła na wniosek i głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości Rada Miasta Puławy. Zygmunta Berlinga nie podlegała polskiemu rządowi na uchodźstwie, ale dowództwu sowieckiemu i realizowała sowiecką rację stanu. Radni wskazywali ponadto, że w pobliżu pomnika w przeszłości funkcjonowała siedziba powiatowego urzędu bezpieczeństwa publicznego, gdzie mordowano polskich patriotów, i z szacunku dla nich pomnik powinien być usunięty. Pomimo usilnych starań sprawa usunięcia pomnika przedłużała się, przede wszystkim ze względu na pat proceduralny związany z nieprzyznawaniem się nikogo do gruntu, na którym był postawiony pomnik. Przełom nastąpił dopiero po przyjęciu ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W uzasadnieniu tej ustawy pomnik w Puławach wymieniono jako jeden z 13 przykładów obiektów, z grupy kilkuset w skali kraju, spełniających kryteria ustawy, który jako symbol totalitarnego systemu winien być usunięty. Ostatecznie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał decyzję nakazującą usunięcie tego pomnika. 20 marca 2018 r. to ważny dzień dla społeczności Puław i regionu. To dzień symboliczny, stanowiący kolejny krok na drodze prowadzącej do zerwania z niechlubną przeszłością. Pomniki na polskiej ziemi mają być i będą stawiane bohaterom i niech tak będzie w Puławach, niech to wolne wreszcie miejsce stanie się miejscem, które uczci patriotów, tych, którzy przelali krew dla wolnej, niepodległej, dumnej Rzeczypospolitej.

16 marca na cmentarzu w Szumowie miałam okazję oddać hołd bohaterom wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Po blisko 100 latach do grobu żołnierzy 201. Ochotniczego Pułku Piechoty w Szumowie trafiły szczątki 10 żołnierzy tego pułku odkryte jesienią zeszłego roku pod Andrzejewem. Stało to się możliwe dzięki inicjatywie Fundacji „Honor, Ojczyzna” i Stowarzyszeniu „Wizna 1939” oraz zaangażowaniu władz gmin Andrzejewo i Szumowo. Ochotniczy Pułk Piechoty? Postawienie tamy bolszewickiej nawale zdawało się zadaniem ponad siły dopiero odradzającej się polskiej armii. Polscy patrioci tłumnie odpowiedzieli na wezwanie ojczyzny i gen. Józef Haller wydał rozkaz o sformułowaniu dywizji ochotniczej. Tych 10 zamordowanych żołnierzy było właściwie jeszcze chłopcami, najstarszy z nich miał 25 czy 30 lat. Wiem to na podstawie przeprowadzanych badań antropologicznych. Byli to harcerze, uczniowie, studenci - przyszłość naszej ojczyzny, którzy bez wahania poświęcili życie, ochraniając odwrót swego pułku w bitwie pod Pęchratką i Paprocią. Powiedziałam, że zostali zamordowani, to nie było przejęzyczenie. Oni nie polegli w walce. Podczas ekshumacji potwierdzono przekazy miejscowej ludności, że jeden z naszych żołnierzy został dobity strzałem w tył głowy, a pozostałym bolszewicy je ścieli. Z perspektywy wojny polsko-sowieckiej śmierć tych 10 chłopców wydawać się mogła tylko nieznaczącym epizodem, w rzeczywistości jednak potwierdza to, z jak strasznym zagrożeniem mieliśmy wtedy do Dzięki bohaterstwu naszych przodków Europy nie zalała fala komunizmu. My, Polacy, podchodzimy do historii na swój wyjątkowy sposób. Wiemy, co zawdzięczamy naszym przodkom, i co im jesteśmy winni. Pragnę serdecznie podziękować delegacji harcerzy ze Skarżyska-Kamiennej, która przybyła do Szumowa, by pożegnać druha Kazimierz Lecha, 15-letniego młodzieńca z Kamiennej, który zginał w bitwie pod Pęchratką i Paprocią. Wiek jednej z ofiar oszacowano na 15 lat i najprawdopodobniej były to szczątki druha Kazimierza. Dziękuję uczniom ze szkoły podstawowej w Szumowie za wieloletnią opiekę nad mogiłą żołnierzy 201. Ochotniczego Pułku Piechoty, a także wszystkim pocztom sztandarowym szkół uczestniczących w uroczystości. Wysoka Izbo! Gros ochotników 1920 r. było harcerzami lub wywodziło się z harcerstwa. Harcerze odegrali wielką rolę już wcześniej, podczas walk o kształt granic naszej odradzającej się ojczyzny podczas powstania wielkopolskiego, powstań śląskich czy obrony Lwowa, a później w latach okupacji. Nawiązując do roli harcerstwa w historii Polski, pragnę powiedzieć, że 10 marca w Piątnicy odbyła się 25. harcerska wieczornica poświęcona twórcy krzyża harcerskiego ks. dr. harcmistrza Kazimierza Lutosławskiego. Bardzo krzepiące jest to, że do tej zasłużonej organizacji, wychowującej wciąż nowe pokolenia polskich patriotów, tak ochoczo garnie się młodzież. 11 tys. instruktorów, w tym 6 tys. drużynowych, nieustannie pracuje nad wykształceniem odpowiednich wartości w młodych ludziach.

Działalność instruktorów przyniosła i wciąż przynosi nieocenione korzyści naszej ojczyźnie i społeczeństwu. Uważam, że powinni być bardziej doceniani, a władze centralne i samorządowe powinny bardziej wspierać działalność organizacji. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie.